Informuję, że w dniu dzisiejszym odbędą się posiedzenia Komisji: - do Spraw Unii Europejskiej wspólnie z Komisją Spraw Zagranicznych - godz. 13.15, - Kultury i Środków Przekazu - godz. 14, - Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki - godz. 18. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 14. porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 437 i 437-A) Bardzo proszę panią poseł Małgorzatę Janowską o przedstawienie uzasadnienia projektu ustawy. Bardzo proszę. Zapraszam serdecznie. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu wnioskodawców projektu mam przyjemność przedstawić państwu pokrótce założenia i cel wniesionego projektu ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw wraz ze złożoną autopoprawką, druki sejmowe nr 437 i 437-A. W 2018 r. w wyniku nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych utworzony został państwowy fundusz celowy - Fundusz Niskoemisyjnego Transportu. Przepraszam panią poseł bardzo. Posłuchajcie państwo. Obruszamy się, gdy ministrowie rządu stoją tyłem i mają nas w nosie. Gdy pani poseł przedstawia, ja bardzo proszę posłanki i posłów o słuchanie. Bardzo serdecznie proszę. Robię to w sposób grzeczny, miły. Proszę bardzo. Dziękuję również. Jego dysponentem został minister właściwy do spraw energii, a zarządcą - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Fundusz został powołany do finansowania takich zadań jak np. rozbudowa infrastruktury umożliwiającej stosowanie paliw alternatywnych. Utworzenie funduszu miało stanowić odpowiedź na brak systemowego wsparcia dla rozwoju rynku oraz infrastruktury paliw alternatywnych w transporcie przy jednoczesnym zobowiązaniu Polski na poziomie dyrektyw Unii Europejskiej do wspierania rozwoju rynku i infrastruktury niezbędnej do wykorzystania paliw alternatywnych. Przyjęty system dysponowania i zarządzania funduszem przewiduje współdziałanie operacyjne aż trzech podmiotów: ministra klimatu, NFOŚiGW oraz Banku Gospodarstwa Krajowego jako podmiotu obsługującego bankowo fundusz. Dodatkowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami, szczegółowy sposób postępowania w zakresie wyboru projektów oraz wsparcia oraz inne szczegółowe warunki są określone przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia. Projektowana ustawa ma na celu uproszczenie, odbiurokratyzowanie i przyspieszenie finansowania ze środków publicznych rozwoju transportu niskoemisyjnego.

Przeniesienie środków finansowych z funduszu i utworzenie zobowiązania wieloletniego pozwoli na przeniesienie środków pomiędzy oboma zobowiązaniami. Zapewni to jak najefektywniejsze finansowanie projektowych celów środowiskowych. Przychodami zobowiązania wieloletniego będą w szczególności środki zgromadzone na rachunku funduszu na dzień jego likwidacji, jak również przychody pochodzące z dotychczasowych źródeł przychodów funduszu.

Powyższa konstrukcja zapewni sprawniejsze wydatkowanie środków na zadania z zakresu transportu niskoemisyjnego. Włączenie realizacji celów przekształconego funduszu do celów statutowych NFOŚiGW zapewni także zwiększenie efektywności wydatkowania środków publicznych oraz odformalizowanie procedur.

W odniesieniu do konkretnych przepisów zawartych w projekcie ustawy omówię pokrótce część z nich. Zmiany zawarte w art. 1 mają na celu umożliwienie przekształcenia państwowego Funduszu Niskoemisyjnego Transportu w zobowiązanie wieloletnie w ramach NFOŚiGW poprzez uchylenie w ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych przepisów dotyczących tego funduszu.

Art. 4 określa dotychczasowe przychody funduszu jako przychody powstającego zobowiązania wieloletniego.

Zmiany zawarte w art. 6 mają na celu uwzględnienie w ustawie zmieniającej ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych skutków przekształcenia funduszu w zobowiązanie wieloletnie. Zmiany w zakresie art. 7 są konsekwencją przejęcia przez NFOŚiGW zadania funduszu polegającego na (Dzwonek) dofinansowaniu Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Zmiana zawarta w art. 8 dotyczy uchylenia art. 20 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, który utrzymywał w mocy akt wykonawczy określający kryteria i warunki udzielania wsparcia ze środków funduszu. W projektowanej ustawie wprowadza się także przepisy przejściowe, które regulują m.in. kwestię rozwiązania umów zawartych pomiędzy NFOŚiGW a BGK w zakresie obsługi przekształconego funduszu czy przejęcia przez NFOŚiGW należności i zobowiązań przekształconego funduszu. Zgodnie z art. 15 przepisy dotyczące wygaszania funkcjonowania funduszu powinny wejść w życie z dniem 30 września 2019 r., natomiast pozostałe zmiany - z dniem 1 października 2020 r. Do pierwotnego brzmienia projektu została dołączona również autopoprawka wprowadzająca zmiany w zakresie art. 4 projektu, czyli ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Dodane w autopoprawce przepisy przyznają właścicielowi jednocześnie sieci przesyłowej i sieci dystrybucyjnej, instalacji magazynowych lub instalacji skroplonego gazu ziemnego albo sieci przesyłowej i sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej uprawnienia w postaci prawa wyboru, czy swoje zadanie będzie realizować jako operator systemu połączeniowego. Autopoprawka ta ma na celu ułatwienie funkcjonowania operatora systemu przesyłowego gazowego w obszarze niskoemisyjnego transportu. Podsumowując, wdrożenie procedur i zasad stosowanych przez NFOŚiGW umożliwi szybsze i efektywniejsze wydatkowanie środków i powiązanie ich z mechanizmami przyjaznymi dla biznesu. Proponowane rozwiązania przyczynią się do wdrożenia programów wspierających rozwój nowoczesnej, innowacyjnej gałęzi gospodarki opartej na elektromobilności. Inwestycje w tym zakresie zapewnią znaczący rozwój sektora przemysłu i usług związanych z transportem niskoemisyjnym, zwiększając także popyt na pojazdy elektryczne, który obecnie jest limitowany ograniczeniami technicznymi, takimi jak niewielki zasięg, wysoka cena oraz niewystarczająca sieć infrastruktury do ładowania. W imieniu wnioskodawców proszę państwa posłów o poparcie przedłożonego projektu. Dziękuję, pani poseł. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Pierwszy poseł, którego proszę, to pan poseł Wiesław Krajewski z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Panie pośle, mam do pana grzeczną prośbę. Wie pan, o co chodzi - żeby wspólnie zrobić coś dobrego. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dziękuję za korektę. Chociaż mam przygotowany materiał, będę się starał przedstawić go w skróconej wersji. W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, zawartego w druku sejmowym nr 437, wraz z autopoprawką, druk nr 437-A. Proponowane zmiany w przedłożonym projekcie ustawy mają na celu przekształcenie państwowego funduszu celowego, Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, w zobowiązanie wieloletnie funduszu w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez uchylenie przepisów dotyczących tego funduszu celowego. W wyniku przekształcenia opłata zastępcza będzie wpływać na rachunek bankowy zobowiązania wieloletniego Funduszu Niskoemisyjnego Transportu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Proponowane zmiany dotyczą m.in. usunięcia z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnienia z opodatkowania podatkiem PIT wsparcia udzielonego ze środków przekształconego funduszu celowego. Zmiany dotyczą również objęcia zwolnieniem z opodatkowania podatkiem CIT dofinansowania udzielonego w formie bezzwrotnej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach zobowiązania wieloletniego. Kolejnym obszarem zmian zaproponowanych przez wnioskodawców są zmiany do ustawy - Prawo ochrony środowiska. Zmiany te mają na celu ujęcie opłaty emisyjnej dotychczasowego funduszu celowego jako przychodu zobowiązania wieloletniego, utworzenie nowego zobowiązania wieloletniego ze wskazaniem celów analogicznych do celów poprzedniego funduszu celowego, skorygowanie odesłań w konsekwencji utworzonego nowego zobowiązania wieloletniego funduszu.

W projekcie ustawy wprowadza się przepisy przejściowe mające na celu nadanie formy prawnej przekształceniu funduszu celowego w zobowiązanie wieloletnie funduszu oraz wskazujące skutki tego przekształcenia w zakresie inwentaryzacji, zamknięcia rachunku, ksiąg rachunkowych oraz sprawozdawczości. Uzupełnieniem omawianych zmian jest autopoprawka wnioskodawców, druk nr 437-A, zmieniająca przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Regulowane zagadnienia mają charakter krajowy i dotyczą kwestii organizacyjnych. Wprowadzone usprawnienia zwiększają dostępność środków dla przedsiębiorców i będą pozytywnie oddziaływać na konkurencyjność gospodarki i rozwój przedsiębiorczości. Wysoka Izbo! Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość rekomenduje przedłożony poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, zawarty w druku sejmowym nr 437, wraz z autopoprawką, druk nr 437-A, i wnosi o jego uchwalenie. Dziękuję, panie pośle. Dziękuję. Posłowie i posłanki PiS-u sprawdzają się co chwilę. Zapraszam panią poseł Urszulę Zielińską, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Szanowni Państwo! Powstanie programu wsparcia niskoemisyjnego transportu rząd ogłosił już w 2016 r. i dzisiejsza dyskusja nad bieżącym projektem jest dobrym momentem, żeby ten program podsumować. O ile rząd ogłosił ten program w 2016 r., o tyle właściwa ustawa umożliwiająca stworzenie Funduszu Niskoemisyjnego Transportu weszła w życie dopiero w połowie roku 2018, a rozporządzenie do tego projektu weszło w życie dopiero pod koniec roku 2019, czyli de facto ten projekt i ten fundusz ruszyły z miejsca dopiero pod koniec zeszłego roku. Fundusz Niskoemisyjnego Transportu miał finansować projekty związane z elektromobilnością, dopłaty do aut elektrycznych, rozbudowę infrastruktury doładowania i tankowania paliw alternatywnych.

Na początku tego roku z mediów dowiedzieliśmy się, że na koncie funduszu jest 360 mln zł, a następnie na czerwcowym posiedzeniu komisji energii dowiedzieliśmy się, że rząd likwiduje fundusz, ale za to uruchamia trzy nowe programy dopłat do aut elektrycznych: „Zielony samochód”, „eVan” i „Koliber”, z tym że na kwotę 147 mln zł, czyli zaledwie 1/5 tego, co przeznaczono, ale nie wydano, na fundusz w poprzednim roku.

Jednocześnie przy każdej kolejnej odsłonie projektu te mniejsze programy, na coraz niższe kwoty, ogłaszane są jako nowe sukcesy i nieważne, że w poprzedniej wersji nie zrealizowano nic, a budżet ucięto lub przesunięto. Co się stało z tymi pieniędzmi? Natomiast co wiemy? Pod tym względem jesteśmy na trzecim miejscu w Europie, ale od końca. Miały być stacje doładowania, jest ich niecałe 1200 sztuk. Pod tym względem jesteśmy na czwartym miejscu w Europie, również od końca.

I wreszcie miało być obniżenie emisji z transportu.

Tymczasem emisje z transportu wzrosły w tym okresie o 80%. To są dane za rok 2018, najnowsze.

Kto więc zyskał na programie? Chyba nikt, może z wyjątkiem tych, którzy zarządzali funduszem, ale tak naprawdę tego też nie wiemy. Podsumowując, chyba można powiedzieć, że program poniósł całkowite fiasko. I dziś tą nowelizacją państwo to przyznajecie. Program nie zadziałał i potrzebuje zmiany, to jest jak najbardziej zrozumiałe, ale ta zmiana powinna być poprzedzona rzetelną analizą tego, co nie zadziałało w poprzednim programie, rozliczeniem wydatków, konsultacją z ekspertami, stroną społeczną. Czy proponowanie tak poważnych zmian w programie, który już raz poniósł tak spektakularne fiasko, bez analizy, bez dyskusji, w trybie ekspresowym to odpowiedzialny plan? Czy może jest to próba wycofania się rakiem z programu, odebrania mu priorytetu, obcięcia środków, rozmycia ich pomiędzy wieloma programami funduszu NFOŚ? Mam nadzieję, że nie, bo też bardzo zależy mi na redukcji emisji, zwłaszcza wysokich emisji z transportu. A czas płynie, panie ministrze, emisje rosną, trujemy dzieci, na ulicach śmierdzi i huczy. A więc aby móc poprzeć ten projekt, [[Dzwonek]] musimy zobaczyć rzetelną analizę wniosków z przeszłości i nowy, przekonujący plan. Będziemy również składać wniosek do biura analiz, aby pomogło w zrozumieniu, co nie zadziałało w tej poprzedniej wersji programu. Dziękuję, pani poseł. Zapraszam pana posła Marka Dyducha, klub parlamentarny Lewica. Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Została przyjęta, bo była taka dyrektywa Unii Europejskiej.

Następnie przyszedł rząd Donalda Tuska, tego Donalda Tuska, który później był twarzą Unii Europejskiej. No mamy ustawę. Następnie przychodzi rząd PiS-u i w 2016 r. pytają tam, w tej Unii Europejskiej: Co wy robicie w kontekście niskoemisyjnego transportu? Mamy ustawę i program. Mamy ustawę, program i fundusz.

Ale jak on miałby funkcjonować, skoro dysponentem w tym ministerstwie był minister środowiska, zarządzającym - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, po drodze był jeszcze minister energetyki, a finanse trzymał Bank Gospodarstwa Krajowego, który się cieszył, bo miał na koncie pieniądze i mógł sobie nimi obracać? Tylko co z tego mieli ludzie? Co one z tego miały?

No to jak wspierały? Przecież oszukiwaliśmy tych ludzi. Oszukiwaliśmy instytucje, oszukiwaliśmy siebie, oszukiwaliśmy Unię Europejską. To jest niestety fakt. Ale teraz zmieniamy ustawę, zmieniamy dysponenta funduszu. To ciekawa sytuacja. Zmieniamy tutaj pięć ustaw, w tym ustawę o podatku od osób fizycznych, ustawę o podatku od osób prawnych, ustawę Prawo ochrony środowiska, ustawę Prawo energetyczne. Poważne ustawy. Tacy zdolni posłowie.

Możemy się założyć w tej sprawie. Co to jest, że posłowie to robią, a nie.

Ale po co się pytać? Jak wnoszą posłowie, to nie ma konsultacji społecznych. W tak ważnej sprawie nie ma konsultacji społecznych. To jest przemądrzały rząd. Bo każdy mądry wie, że jak jest duży problem, to trzeba uruchomić inicjatywę, trzeba uruchomić mobilność tych ludzi i ich umysły. Dlaczego my mamy kupować technologię - bo tak to się skończy, że będziemy kupować za te pieniądze technologię - zamiast ją sprzedawać? Co, Polacy są głupsi od innych narodów? Można byłoby to wykorzystać, a my przerzucamy. I teraz - ostatnie słowo: fundusz. Te pieniądze idą do narodowego funduszu ochrony środowiska. To świetnie, tylko że narodowy fundusz ochrony środowiska w innych dziedzinach wydaje ok. 50% środków. Ja nie widzę tu gwarancji.

Mamy nadzieję, że rząd je po prostu wykorzysta. Dziękuję serdecznie.

Chciałbym bardzo też serdecznie podziękować koleżankom i kolegom, którzy z jednej strony... i pani sprawozdawcy projektu, jak również tym, którzy zabierali głos przede mną, bo część argumentacji została, że tak powiem, już przedstawiona.

Tak to odczuwam, że de facto jest to projekt rządowy. Powołuje się zobowiązanie wieloletnie Fundusz Niskoemisyjnego Transportu w narodowym funduszu ochrony środowiska. Zmienia się również tego, kto dysponuje tym kontem.

De facto to jest główne źródło finansowania tego funduszu. Czemu ma służyć ta nowela?

Brak jest jasnych przesłanek, co ma poprawić ta zmiana prawa w zakresie efektów rozwoju niskoemisyjnego transportu. Zmienia się ustawowe zobowiązania na cele ustalone przez Radę Nadzorczą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest pytanie, czy ustawodawca chce świadomie rezygnować z tego, żeby akurat grono, jakim jest rada nadzorcza, określało te cele, które miały stanowić jedną z podstaw rozwoju i modernizacji tego sektora transportu. Nic nie mówi się o wysokości środków gromadzonych i zmianach po wprowadzeniu zobowiązania wieloletniego. Fundusz Niskoemisyjnego Transportu ulega likwidacji przed uruchomieniem jakichkolwiek działań w zakresie transportu, a w tym celu był stworzony. Powinniśmy ocenić, dlaczego tak się dzieje, jakie są tutaj punkty oporu, które sprawiają, że działa on nieefektywnie, jak sądzę, bo chyba stąd ta zmiana. Był on przyczynkiem do ustanowienia opłaty zastępczej, narodowego celu wskaźnikowego, czyli zamiany obniżenia ilości biokomponentów i biopaliw na rynku ustalonego na dany rok za tę opłatę, przy czym ta opłata de facto jest 10 razy niższa niż koszt zakupu biokomponentów, czyli odbywa się to kosztem rozwoju sektora biopaliw, również rolników, którzy produkują surowce rolnicze potrzebne dla tego rozwoju. Jak będą rozdysponowane? Pytanie o równomierne traktowanie również poszczególnych technologii w zakresie rozwoju niskoemisyjnego transportu, czy sektor biopaliw utrzyma tam swoje należne miejsce, czy tylko będzie preferowana elektromobilność, czy w tworzeniu funduszu celowego będzie mógł ten sektor biopaliw liczyć również na odpowiednie wsparcie. W większości krajów, przynajmniej w połowie krajów Unii Europejskiej, taki produkt już wdrożono. Wdrożenie takiego produktu wymaga edukacji i promocji. Rozporządzenie wykonawcze do Funduszu Niskoemisyjnego Transportu wydane przez ministra do spraw energii zakładało promocję etyliny 10. Czy znajdzie to uznanie w kierunkach ustalanych przez Radę Nadzorczą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej? Nie mamy na to odpowiedzi. Nowelizacja ogranicza do zera do roku 2027 wydatki z budżetu związane z kierunkami rozwoju, jakie miał wspierać likwidowany Fundusz Niskoemisyjnego Transportu. Pytanie: Dlaczego? Branża biopaliw, branża rolnicza bardzo ostro protestowała przy ostatniej nowelizacji ustawy, gdzie wprowadzono narodowy, gdzie narodowy cel wskaźnikowy był redukowany opłatą zastępczą, i w chwili obecnej ma też taki dylemat. O to bardzo trudno było w dyrektywie RED II o odnawialnych źródłach energii. Ochronić 7-procentowy udział biopaliw z surowców rolniczych do roku 2030, a jednocześnie mamy do roku 2030 14% udziału OZE w transporcie i ten cel jest poza zasięgiem, jeżeli nie wykorzystamy akurat tych (Dzwonek) 7% udziału biopaliw z surowców rolniczych, nie mówiąc o tym, co to daje dla sektora rolniczego. To są pasze, to jest płodozmian, to jest wiele innych celów. Tak że ta zmiana to nie tylko pięć ustaw wskazanych w tej ustawie, ale również konsekwencje, które mogą dotyczyć wielu różnych sektorów, i na to chciałem zwrócić uwagę. Nie sprzeciwiamy się przekazaniu tego do komisji, ale uważamy, że na te pytania powinniśmy uzyskać odpowiedź w trakcie prac w komisji. Dziękuję za ten mądry, rozsądny, fajny głos, panie pośle. Miło się słuchało. Pan poseł Dobromir Sośnierz jest proszony na mównicę, Koło Poselskie Konfederacja. Witam pana, panie pośle. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Na początek chciałbym się trochę nie zgodzić z kolegami przedmówcami, z panem Markiem Dyduchem i panem Andrzejem Grzybem.

Jeśli problemem jest to, że nie ma konsultacji społecznych, to wprowadźmy konsultacje społeczne dla projektów poselskich - i to jest rozwiązanie, a nie to, że rząd pisze ustawy. Ale wracając do rzeczy, socjalizm jest to taki ustrój, który bohatersko rozwiązuje trudności, które wcześniej sam stwarza, i dokładnie tak jest w tym przypadku. Najpierw powołujemy dodatkowy Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, a po 2 latach orientujemy się, że niepotrzebnie, bo to samo, ba, nawet lepiej, można by rozwiązać bez tego funduszu w ramach już istniejących instytucji. No i tak brniemy od sukcesu do sukcesu, cytując pana Michalkiewicza. Za każdym razem mamy powody do radości, najpierw powołujemy fundusz z oklaskami, później oklaski, że go odwołujemy. Znając życie, to zresztą niekoniecznie jakieś mądre powody muszą stać za tym wnioskiem, że ten fundusz nam jest niepotrzebny. Być może przecież jest tak, jak to w praktyce rządów naszej neosanacji bywa, że po prostu osoba, dla której ten fundusz utworzono, żeby miała gdzie pracować, okazała się niewdzięcznikiem albo z innych powodów stała się zbędna i teraz fundusz likwidujemy. Ale nie wiem, może jednak są inne powody. Ale problem polega na tym, że ten wniosek, że nie potrzebujemy tego funduszu, jest po prostu nie dość daleko idący, bo nie tylko nie potrzebujemy tego funduszu, lecz także po prostu nie potrzebujemy tego, żeby państwo, żeby urzędnicy decydowali, jaka technologia jest nowoczesna, innowacyjna czy przyszłościowa, a jaka nie jest. Jeśli technologia jest przyszłościowa, to przyszłość nam to pokaże - i nie potrzebujemy do tego urzędników do odgadywania przyszłości. Z historii zresztą znamy wiele przypadków, jak to urzędnicy próbowali zadekretować przyszłość i angażowali pieniądze podatników w różne projekty, które dzisiaj raczej budzą rozbawienie. Pod koniec XIX w. rządy wzywały tęgie głowy na obrady, jak rozwiązać problem zalegających w miastach końskich odchodów w związku z szybkim rozwojem transportu miejskiego. Prognozowano, że jak tak dalej pójdzie, to końska kupa będzie niedługo zasłaniać ludziom widok z drugiego piętra. Organizowano w tej sprawie takie odpowiedniki naszych dzisiejszych szczytów klimatycznych, podczas których tęgie głowy radziły nad tym bez końca i - dokładnie tak jak na naszych współczesnych szczytach klimatycznych - nie potrafiły wyjść poza ekstrapolację tego, co już znają. Problem by się nie rozwiązał, gdyby nie to, że jakiś prywaciarz wynalazł samochód i całe te dywagacje stały się zbędne. Ale państwa początkowo wcale nie odnosiły się do tego projektu z entuzjazmem, do samochodów. W dalekim mieście Warszawa ponoć nadal rządzi człowiek, który próbuje zwalczać samochody, i nawet próbowano zakazywać wjazdu do miast samochodów, ulegano lobbingowi woźniców, którzy protestowali przeciwko tej nieuczciwej konkurencji. Tak było. Warto też pamiętać, że niektóre rządy za słuszną technologię jeszcze nie tak dawno uważały diesla, stosowały różne zachęty finansowe, programy rozwojowe, żeby do diesla zachęcać, po czym w którymś momencie uznały, że jednak diesel jest zły, i zaczęły go prześladować, zwalczać, zakazywać wjazdu do centrów miast, wystawiając do wiatru tych, których wcześniej do tego zachęcali, którzy tych zachęt rządowych wcześniej słuchali. Teraz się okazuje, że restrykcje wobec diesli też były raczej pochopne, niepotrzebne i wcale nie przynoszą oczekiwanych efektów. To pokazuje, jak kiepsko urzędnicy i finansowane przez nich projekty są w stanie odgadywać tę przyszłość. Te przykłady powinny nas nauczyć więcej pokory w stosunku do pomysłów urzędników na rozwój techniki. Rządy wielokrotnie ładowały pieniądze podatników w nieudane projekty albo zwalczały technologie, które potem okazywały się rzeczywiście przyszłościowe. Urzędnicy oprócz tego bowiem, że się mylą po prostu po ludzku, wydają się też niestety podatni na tzw. pozamerytoryczne środki przekonywania, czyli po prostu na korupcję ze strony lobbystów promujących różną technologię. A więc dużo lepiej, myślę, zrobimy, jeśli urzędnicy przestaną się po prostu mieszać w rozwój techniki i zostawią to rynkowi.

Zastanówcie się, jaka jest szansa, że tutaj ta nasza technologiczna pustynia wyda jakiś urodzajny owoc w tej dziedzinie, na rynku, na którym nie mamy do tej pory żadnych istotnych osiągnięć. Żeby to miało sens, to musi najpierw tu powstać przemysł, który nadgoni te zaległości. Żeby taki przemysł powstał, muszą istnieć po prostu liberalne, sensowne przepisy gospodarcze i takie przekonanie, zaufanie ze strony inwestorów, że państwo jest stabilne, a nie np. wypluwa z Sejmu ustawy w takim tempie, że posłowie nie nadążają z czytaniem. W takim kraju nikt nie będzie chciał inwestować. Oczywiście pod warunkiem, że ona jest sensowna, a póki co wiele wskazuje na to, że niestety nie jest. Gdyby auta elektryczne były dobre, to ludzie sami by je kupowali, nie trzeba by ich do tego zachęcać, a póki co ładujemy pieniądze jednych podatników w to, żeby drudzy kupili sobie nowe auto, i to często pieniądze tych, których nie stać na nowe auto.

Dziękuję, panie pośle. Proszę państwa, przechodzimy do pytań. Ustalam limit czasu na 1 minutę. Zapraszam pana posła Mirosława Suchonia z Koalicji Obywatelskiej. W związku z tym zapraszam pana posła Pawła Krutula z klubu parlamentarnego Lewica. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przedłożony projekt zakłada utworzenie Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, którego celem jest finansowanie rozbudowy infrastruktury umożliwiającej stosowanie paliw alternatywnych, w tym biokomponentów. W ramach tego projektu realizowany jest program wsparcia w zakupie samochodów dostawczych z napędem elektrycznym.

Liczba samochodów objętych dofinansowaniem wynosi 1 tys. sztuk. Według portalu Wysokie Napięcie wnioski o zakup aut złożyło do tej pory zaledwie dziewięciu przedsiębiorców. Moje pytanie brzmi: Kiedy i czy ministerstwo planuje wprowadzenie programu realnie zachęcającego do zakupu pojazdów z napędem elektrycznym? Dziękuję serdecznie. Zapraszam pana posła Marka Rutkę, klub parlamentarny Lewica. Wasza Marszałkowość! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Obecnie w Polsce zarejestrowanych jest nieco ponad 8 tys. samochodów z napędem elektrycznym, z czego auta w pełni elektryczne stanowią zaledwie 59%. Resztę stanowią auta typu plug-in. Warto wspomnieć, że zgodnie z założeniami dokumentu pn. „Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych” autorstwa Ministerstwa Energii w 2017 r. zakładano, że w 2020 r. na polskie drogi wyjedzie ponad 44 tys. samochodów z napędem elektrycznym, a w 2025 r. będzie ich ponad 1 mln. Tak więc w takim tempie na obiecywany przez premiera Mateusza Morawieckiego 1 mln aut elektrycznych przyjdzie nam czekać 125 lat. Moje pytanie brzmi: Czy ministerstwo może zagwarantować, że wielkość 1 mln aut elektrycznych osiągniemy trochę szybciej niż w 2145 r., czyli np. do roku 2030?

Dziękuję serdecznie waszej posłowości. Zapraszam pana posła Krzysztofa Gadowskiego z Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska, znanego z tego, że lubi sobie pogadać przez telefon głośno, tak że wszyscy słyszymy. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Miał być fundusz, który miał przyczynić się do rozwoju elektromobilności, miała powstać do tego infrastruktura. Dlatego, panie ministrze, pytam: Jaka jest dzisiaj wartość tego funduszu? Kiedy faktycznie pierwsze pieniądze z tego funduszu wydano na zadania określone w zapisach statutu tego funduszu? Jakie państwo poniosło koszty, społeczeństwo polskie, na administrację, funkcjonowanie tego funduszu? Co prawda one były podane, wyspecyfikowane w ustawie w 2018 r. Czy ta nowa formuła, którą wprowadzacie, poprawiając działanie Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, przyczyni się [[Dzwonek]] do sprawniejszego wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na konkretny cel zapisany w statucie i misję tego funduszu? Dziękuję serdecznie. Zapraszam.

Celem tego funduszu powołanego 2 lata temu było zmniejszenie emisyjności właśnie spalin pochodzących z benzyny, pochodzących z oleju napędowego. W ciągu 2 lat od powołania tego funduszu dokładnie nic nie zrobiono. Samorządy w ramach posiadanych środków robią to, co mogą. Chciałam zadać pytanie w związku z zapowiedziami w tej zmienianej kolejny raz ustawie, bo ona pochodzi z 2006 r. i przez 14 lat niewiele w tej sprawie zrobiono.

Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Zapraszam. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Fundusz Niskoemisyjnego Transportu miał być głównym źródłem finansowania rozwoju elektromobilności w Polsce. Szumnie zapowiadano rozdysponowanie na różne projekty prawie 7 mld zł. Pytam: Gdzie te samochody elektryczne obiecane przez premiera Morawieckiego? Dla samorządów kluczowy jest nie tyle sposób gromadzenia środków na poziomie centralnym na potrzeby udzielania wsparcia finansowego, co sprawne i przejrzyste działanie. Jest to o tyle ważne, że nałożyliście na samorządy szereg obowiązków, którym muszą podołać, np. zapewnienie udziału co najmniej 30% pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów. Pytam zatem: Dlaczego ten projekt został zgłoszony jako projekt (Dzwonek) poselski, bez żadnej współpracy z samorządami, np. w ramach prac Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego? Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. A teraz pytanie, na które czekam ze szczególnym zainteresowaniem. Pan poseł Janusz Korwin-Mikke. Będziemy się łączyli. Ja chciałem tylko spytać, czy obecni na sali zdają sobie sprawę, że zabierają głos na temat, na którym się w ogóle nie znają. Gdyby 125 lat temu Kongres amerykański zajął się problemem rozwoju motoryzacji, zajął się problemem zapewnienia paliwa dla powstających samochodów i uruchomił specjalny fundusz, który pomoże przedsiębiorcom, i drugi fundusz, który pomoże producentom paliw, gdyby jeszcze rząd amerykański skonsultował to z organizacją państw amerykańskich, a nie daj Boże, jeszcze zrobił konsultacje społeczne, to do dzisiaj jeździlibyśmy konno, bo, jak słusznie zauważył śp. Henryk Ford: gdybym spytał ludzi, czego potrzebują, powiedzieliby, że potrzebują większych, szybszych i tańszych koni.

A teraz jest nawet nie to, co my chcemy, tylko tyle, ile powstaje z tego potworka, jakim są ustawy. Dziękujemy serdecznie, panie pośle. Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Fundusz na niskoemisyjny transport to jest najbardziej tajemnicza ustawa 14. posiedzenia Sejmu.

I teraz należy zadać sobie pytanie: O co tu tak naprawdę chodzi?

Niemniej po prostu mamy do czynienia z jakimiś bardzo dziwnymi ruchami.

I ostatnia uwaga, jeśli pan marszałek szanowny pozwoli, z którą, mam nadzieję, pan marszałek. Oboje jesteśmy posłami ze Śląska. Tam kwestie zanieczyszczenia, kwestie ekologiczne są szczególnie ważne. I z tego punktu widzenia tak ważne jest, żeby te pieniądze zostały jak najszybciej w najlepszy sposób spożytkowane na transport niskoemisyjny i po drodze nigdzie nie zginęły. Ja co prawda jestem posłem z Zagłębia, ale generalnie mniej więcej tamten kierunek. Pan poseł Stefan Krajewski, zapraszam serdecznie, klub parlamentarny PSL - Kukiz15, Koalicja Polska oczywiście. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Już się przyzwyczailiśmy do tego, że rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd Zjednoczonej Prawicy kugluje - kugluje pieniędzmi, kugluje zadaniami, łączy instytucje, dzieli. Dzisiaj widzimy, że będzie likwidowany fundusz celowy, po to żeby pieniądze, żeby zadania przenieść do dużego narodowego funduszu ochrony środowiska. Nie będzie widać, ile pieniędzy wydane, na jakie cele, łatwiej przesuwać te pieniądze. Była obietnica miliona aut elektrycznych. Mamy milion pojazdów, pewnie więcej, ale tylko hulajnogi mamy niestety, a nie samochody. Orlen wszystko jest w stanie lepiej zrobić, hot-dogi Lotosu będzie sprzedawał teraz z logo Orlenu i już będzie pełen sukces tego rządu. A więc i to mógłby też wykorzystać, mógłby to robić. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Zapraszam pana posła Grzegorza Brauna z Konfederacji, klubu parlamentarnego... koła, koła. Ale życzę wam klubu kiedyś oczywiście. Klub to przyszłość, mam nadzieję, niedaleka. Zapraszamy - zapraszamy do Konfederacji. Szanowni państwo, jeśli staracie się tutaj wyczuwać trendy przyszłości, to właśnie my. Wysoka Izbo! Moje pytanie: Co o tym wszystkim sądzi pan premier, który osobiście zaangażował swój autorytet indywidualny, a także majestat Rzeczypospolitej, w ten projekt?

Przelewacie pieniądze z pustego w próżne do innego urządzenia do mielenia pieniędzy, które się wcześniej odebrało podatnikom. Co o tym sądzi pan premier? Bo jeżeli wcześniej tak się angażował, a teraz państwo podejmujecie decyzję o kasacji, o zezłomowaniu tego waszego Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (Dzwonek), to może pan premier wie o czymś ważnym, co o tym przesądza. No i konkretnie, czy może kontynuując światłą myśl moich znakomitych kolegów: Sośnierza i Korwina, może trzeba już rozglądać się za jakimś wierzchowcem, bo jeżeli to jest tendencja regresywna i jeżeli z elektrycznych aut nic nie będzie, to może i nieelektryczne trzeba będzie niedługo zezłomować i może wobec tego. Co sądzi o tym pan premier? Konkretne pytanie. Skoro panu premierowi. Dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie za to błyskotliwe pytanie. Zapomniał pan zresztą o swoim tradycyjnym: Szczęść Boże, czym złamał pan moje serce. Zapraszam, panie pośle. Niech pan się tak nie spieszy, nie uciekniemy panu. Jest. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam dwa pytania w związku z tym projektem ustawy.

Dziękuję bardzo. Zapraszam pana posła Franciszka Sterczewskiego z Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska. Panie pośle, mównica jest pana. Wysoka Izbo! Panie Ministrze!

To jest skandal. To jest skala wstydu naszego rządu. Dlaczego zatem likwiduje się Fundusz Niskoemisyjnego Transportu? Czy rząd planuje jakiś program dofinansowań dla obywateli i obywatelek np. na zakup rowerów [[Dzwonek]] elektrycznych, które są dużo bardziej potrzebne niż samochody? Dziękuję serdecznie.

Najpierw spieszę z wyjaśnieniem panu posłowi Sośnierzowi, że nie jestem przeciwko inicjatywie poselskiej. Powiedziałem tylko w ten sposób, że ta zmiana ustawy nosi wszelkie znamiona projektu rządowego, tylko że była złożona przez posłów. Tylko tyle. Natomiast chciałbym drążyć kwestię opłaty zastępczej pochodzącej w dużej mierze z sektora biopaliw, bo ona de facto redukuje ilość wytwarzanych czy wprowadzanych na rynek biokomponentów i biopaliw. I tutaj, proszę państwa, chciałbym na tej sali powiedzieć: ogromną zasługę, jeśli chodzi o ochronę 7-procentowego udziału biopaliw pochodzących z surowców rolniczych, ma m.in. Krajowa Izba Biopaliw. Bardzo żałuję, że tego podmiotu nie doceniamy przy noweli tej ustawy. Bez ich determinacji.

Bez ich udziału, bez ich determinacji naprawdę nie mielibyśmy tego 7-procentowego udziału.

Dziękujemy serdecznie za podniesienie tej kwestii.

Panie ministrze, ma pan 5 minut. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Bardzo się cieszę z wielkiego zainteresowania tym projektem, bo to jest rzeczywiście ważny kierunek rozwoju naszego kraju, ważny kierunek, jeśli chodzi o poprawę jakości powietrza w Polsce.

Proszę państwa, mówię do posłów Platformy Obywatelskiej. Była o to awantura. Uprzejmie proszę: jak mówi minister, słuchają posłowie. Panie ministrze, ma pan głos. Odnosząc się do kilku konkretnych uwag, które były adresowane do rządu w waszych wypowiedziach, mogę zagwarantować, że wszystkie te środki, które zostaną właśnie przeniesione z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu do narodowego funduszu, zostaną przeznaczone na dokładnie takie same cele. Tak brzmi właśnie ta propozycja - żeby wykorzystać te środki dokładnie na te same cele.

Wydaje mi się, że to tyle, jeśli chodzi właśnie o te konkretne pytania, które były adresowane do nas. Proszę państwa, zamykam dyskusję. Marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu, proponuje, aby Sejm skierował poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, zawarty w drukach nr 437 i 437-A, do Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych w celu rozpatrzenia. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Proszę państwa, pół minuty przerwy i przechodzimy do spotkania z naszą kochaną panią marszałek Witek. Dziękuję serdecznie.

Wznawiam obrady. Bardzo proszę wszystkich państwa posłów o naciśnięcie dowolnego przycisku w celu stwierdzenia kworum. Bardzo proszę.

Stwierdzam kworum. Właściwe komisje przedłożyły sprawozdania o uchwałach Senatu w sprawie ustaw: - o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców, - o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw. Sprawozdania to druki nr 485 i 479. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkty obejmujące rozpatrzenie tych sprawozdań. Proponuję, aby w tych przypadkach Sejm wyraził zgodę na skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Wybraliście mnie państwo na samym początku kadencji członkiem Komisji do Spraw Kontroli Państwowej. Niestety, większość sejmowa odebrała niedawno możliwość zwoływania posiedzenia przewodniczącemu naszej komisji, a sytuacja jest nadzwyczajna i wymaga pilnego, niejawnego spotkania, by wysłuchać prezesa Banasia i otrzymać raport ukazujący obraz ostatnich wydarzeń w Najwyższej Izbie Kontroli. Prezes NIK złożył doniesienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez wiceprezesa NIK, do niedawna posła PiS-u, pana Dziubę i odsunął go od wykonywania obowiązków służbowych. W związku z tym, pani marszałek, zwracam się z wnioskiem formalnym do pani marszałek, bo nie ma innej możliwości, żeby była pani uprzejma zwołać takie tajne, poufne, niejawne posiedzenie naszej komisji.

Proszę bardzo.

Kłaniam. Szczęść Boże! Wysoka Izbo!

Fałszywa pandemia” to zbiór tekstów uczonych, medyków. Czas się ogarnąć, czas przestać straszyć naród, a także posłów restrykcjami związanymi z pewną rozbudowaną, wielopoziomową fikcją polityczno-propagandową. Dziękuję, pani marszałek. Wobec tego nie głosujemy nad tym wnioskiem, Konwentu zbierać nie będę. Powracamy do rozpatrzenia punktu 1. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o wsparciu dla rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 482-A. Proszę pana posła Henryka Kowalczyka o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Do ustawy zgłoszono w czasie drugiego czytania cztery poprawki. Komisja Finansów Publicznych rozpatrzyła w dniu wczorajszym wszystkie poprawki. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 482. Komisja przedstawia w dodatkowym sprawozdaniu poprawki, nad którymi Sejm będzie głosować w pierwszej kolejności.

Sejm poprawkę odrzucił. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 2. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 3. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 4. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm poprawkę przyjął.

Dziękuję pani marszałek, że pozwoliła mi zabrać głos, bo rzecz jest najwyższej sprawy. Chcecie objąć system ubezpieczeń wierzytelności handlowych gwarancjami państwa, tylko że robicie po raz kolejny ten sam błąd. Przed laty wstrzymywaliście państwo, by objęło kontrolą SKOK-i, a jednocześnie SKOK-i zostały objęte gwarancją BFG. Dzisiaj dokładnie to samo chcecie zrobić z zakładami ubezpieczeń, które ubezpieczają wierzytelności handlowe. Tak, rynek się zblokował, to prawda. Trzeba rynkowi pomóc, ale trzeba to zrobić z głową, wprowadzając systemowe rozwiązania ważenia ryzyka, oceny transakcji, weryfikacji rzetelności. Firmy ubezpieczeniowe potrafią naprawdę bardzo różnie pracować.

Nie ma czegoś takiego jak skutki gospodarcze COVID-19. Są skutki waszych decyzji i zaniechań w tej sferze. Są skutki sprowadzania przez was powszechnego niebezpieczeństwa poprzez zamrażanie życia gospodarczego. Tego skutki obserwujemy. Katastrofa społeczno-gospodarcza i nadużycie uprawnień jako główna zasada ustrojowa Rzeczypospolitej trzeciej i pół.

za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 482, wraz z przyjętą poprawką, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm uchwalił ustawę o wsparciu rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19. Wniosek formalny. Proszę bardzo, z wnioskiem formalnym, pani poseł. Szanowna Pani Marszałek! Dla posłów reglamentuje pani ilość miejsc w trakcie posiedzenia Sejmu. Zwracałam się do pani w trakcie posiedzenia, że w ławach poselskich, a nie w ławach rządowych, siedzi wiceminister, nie poseł, wraz z dyrektorem, i prosiłam panią o interwencję. Dobrze, że w tym momencie pani minister się zreflektowała i wyszła. Ale poproszę, żeby pani w przyszłości, tak jak pani próbuje dyscyplinować opozycję, w stosunku do swoich koleżanek i kolegów podobne rygory zachowywała. A w tym przypadku w sposób szczególny, skoro jest przeznaczone na to miejsce. A już sytuacją zadziwiającą jest to, że dyrektor departamentu jednego z ministerstw może zasiadać w ławach rządowych. Pani poseł, prowadząc obrady, nie jestem w stanie rozpoznać, kto jest posłem, a kto nie. Jeżeli jest taka sytuacja. Ale proszę. No po co? Powracamy do rozpatrzenia punktu 2. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 480-A. Przystępujemy do trzeciego czytania. Proszę pana posła Krzysztofa Tchórzewskiego o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji. Wysoki Sejmie! W trakcie drugiego czytania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii złożony został wniosek o odrzucenie projektu ustawy w całości oraz cztery poprawki. Komisja po rozpatrzeniu wniosku i poprawek rekomenduje Wysokiej Izbie głosowanie przeciw wnioskowi o odrzucenie projektu ustawy oraz rekomenduje odrzucenie zgłoszonych poprawek. Komisja przedstawia w dodatkowym sprawozdaniu wniosek o odrzucenie projektu ustawy w całości oraz poprawki. W pierwszej kolejności pod głosowanie poddam zgłoszony w dyskusji wniosek o odrzucenie projektu ustawy. Przyjęcie tego wniosku spowoduje bezprzedmiotowość propozycji komisji. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie projektu ustawy w całości, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm wniosek odrzucił.

Komisja wnosi o ich odrzucenie.

Sejm poprawki odrzucił. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 2. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Stwierdzam, że Sejm poprawkę odrzucił.

Wysoka Izbo! Jest błędem ustrojowym to, że musimy zajmować się specjalną ustawą, żeby uporządkować sprawy Lasów Państwowych. Natomiast przy okazji ustawy o odnawialnych źródłach energii trzeba podnieść jedną fundamentalną kwestię i zadać rządowi jedno fundamentalne pytanie: Jak rząd zamierza obronić Polskę przed agendą nowego zielonego ładu proponowanego w Unii Europejskiej, który będzie niszczył naszą energetykę, będzie sprawiał, że ceny prądu będą rosły, który nie pozwoli na ewolucyjną transformację naszej gospodarki, również sektora energetycznego, tylko będzie służył interesom głównie Niemiec, Francji?

Dziękuję. Szanowni Państwo!

Jeśli państwo pozwolą, drugie pytanie. Czy chcecie uzależnić przedsiębiorstwo Lasy Państwowe od jednego odbiorcy, Skarbu Państwa, który będzie kupował od nas po zawyżonych cenach, rujnując przemysł drzewny w Polsce, i który będzie importował? To jest przepis na zrujnowanie przedsiębiorstwa Lasy Państwowe i uzależnienie go od Skarbu Państwa. Dziękuję, pani poseł.

Wysoka Izbo!

Szanowni Państwo! Zadałem już to pytanie i zadam je dzisiaj: W czyim interesie zaczęliście tak gigantyczną skalę manipulacji? W czyim interesie? Wysoka Izba musi wiedzieć, że polskie elektrownie, polskie elektrownie importują 2,5 mln t biomasy. Skąd importują? Z Czech, z Austrii, z Republiki Federalnej Niemiec, ze Wschodu.

Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projekt ustawy w brzmieniu z druku nr 480, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Propozycją zaopiniowaną przez Prezydium Sejmu jest, aby Sejm skierował projekt ustawy zawarty w druku nr 452 do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w celu rozpatrzenia. W dyskusji zgłoszono wniosek o przystąpienie niezwłocznie do drugiego czytania, bez odsyłania projektu do komisji. Ten wniosek poddam pod głosowanie. Jego odrzucenie będzie oznaczało, że Sejm skierował projekt ustawy do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o przystąpienie niezwłocznie do drugiego czytania projektu ustawy zawartego w druku nr 452, bez odsyłania do komisji, zechce nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił, a tym samym skierował projekt ustawy do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 15. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju o uchwale Senatu w sprawie ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (druki nr 444 i 485) Proszę pana posła Krzysztofa Tchórzewskiego o przedstawienie sprawozdania komisji. Wysoki Sejmie! W imieniu sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju przedstawiam sprawozdanie komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Wysoki Sejmie! Senat zgłosił 45 poprawek do tej ustawy. Komisja Gospodarki i Rozwoju rekomenduje Wysokiej Izbie przyjęcie wszystkich poprawek zgłoszonych przez Senat. Ze względu na współzależność proponujemy także grupowe głosowanie w przypadku niektórych z tych poprawek. To także poparło Biuro Legislacyjne Senatu. W związku z tym zamiast 45 będziemy mieli 9 głosowań. Przypominam, że Sejm odrzuca poprawki Senatu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Jeżeli Sejm nie odrzuci poprawki Senatu, uważa się ją za przyjętą. W punktach porządku dziennego dotyczących rozpatrywania poprawek Senatu głosować będziemy nad wnioskami o odrzucenie poprawek Senatu.

Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie. Komisja wnosi o ich przyjęcie. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem ww. poprawek, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawki przyjął.

Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie.

Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawki przyjął. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 6. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął.

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 21. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął. Głosujemy.

Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawki przyjął.

Głosujemy.

Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawki przyjął.

Komisja wnosi o ich przyjęcie.

Nikt nie był za, przeciw - 449, nikt się nie wstrzymał. Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawki przyjął. Głosujemy.

Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 35. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął. Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Bardzo proszę.

Wznawiam obrady. Proszę państwa, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów podjęłam decyzję o zdjęciu z porządku dziennego trzeciego czytania poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami, druki nr 420, 451 i 451-A. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 16. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (druki nr 447 i 479) Proszę pana posła Bolesława Piechę o przedstawienie sprawozdania komisji. Wysoka Izbo! W imieniu Komisji Zdrowia mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Zdrowia o uchwale Senatu w sprawie zmiany ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw. Komisja 14 lipca rozpatrzyła te poprawki i rekomenduje Wysokiej Izbie z 22 zgłoszonych poprawek przyjąć 15 i odrzucić siedem. Przy czym, w porozumieniu z Biurem Legislacyjnym Sejmu, rządem oraz legislacją Senatu, część poprawek została zblokowana, w związku z tym będziemy mieli do rozstrzygnięcia 15 poprawek. Senat zgłosił do art. 1 ustawy nowelizującej zawierającego zmiany do ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komisja wnosi o ich przyjęcie.

się wstrzymał?

Głosujemy.

1 - za, przeciw - 447, 1 się wstrzymał.

Komisja wnosi o ich przyjęcie. Kto jest przeciw?

Wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów Sejm poprawki przyjął.

Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki.

Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.

Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 7. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Nikt nie był za, przeciw - 449, 1 się wstrzymał. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Głosujemy.

Głosujemy. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 11. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów. Głosujemy.

Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów. Z poprawką tą łączy się 16. poprawka. Głosujemy.

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 15. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 18. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął.

Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawki przyjął. Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw oraz zakończyliśmy głosowania w dniu dzisiejszym. Ogłaszam 5 minut przerwy.

Wznawiam obrady. Przypominam, że postawienie pytania nie może trwać dłużej niż 2 minuty, zaś udzielenie odpowiedzi nie może trwać dłużej niż 5 minut. Prawo do postawienia pytania dodatkowego przysługuje wyłącznie posłowi zadającemu pytanie. Dodatkowe pytanie nie może trwać dłużej niż 1 minutę, a uzupełniająca odpowiedź nie może trwać dłużej niż 3 minuty. Marszałek Sejmu może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu odpowiedzi na pytania dodatkowe. Proszę państwa, rozpoczynamy od pytania pana posła Mieczysława Kasprzaka z klubu parlamentarnego PSL-Kukiz15, Koalicja Polska, w sprawie pomocy dla osób i samorządów poszkodowanych w wyniku lokalnych powodzi. To pytanie będzie zadawane prezesowi Rady Ministrów, w którego imieniu odpowie podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pani minister Anna Moskwa. Udało mi się. Panie pośle, zapraszam serdecznie. Dziękuję, panie marszałku. bo temat jest bardzo trudny i skomplikowany. Pozwoliłem sobie skierować, panie marszałku, zapytanie do pana premiera w zakresie pomocy dla poszkodowanych w czasie powodzi na przełomie czerwca i lipca, które nawiedziły Podkarpacie.

Przybór wód był tak szybki, że niektórzy nie zdążyli ewakuować się ze swoich pomieszczeń.

Potrzebne są pieniądze na odbudowę. Samorządowcy mają wiele uwag do funkcjonowania Wód Polskich, które nie wywiązują się właściwie z konserwacji, z przeglądu cieków wodnych. Dlatego skierowałem do pana premiera pytania, które m.in. kierują do mnie samorządowcy. Kiedy samorządy otrzymają środki finansowe na usuwanie skutków nadmiernych opadów i huraganów? Jakie to będą środki finansowe? Czy państwowe gospodarstwo Wody Polskie podejmie zdecydowane działania, jeżeli chodzi o poprawę stanu rzek i potoków? Kolejne pytanie: Kiedy zostanie opracowane strategiczne rozwiązanie dotyczące gospodarki wodnej, w tym budowy zbiorników retencyjnych? Jest to poważna sprawa. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie pośle. Na pana pytanie spieszy odpowiedzieć pani minister Anna Moskwa. Proszę bardzo. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pozwolę sobie odpowiedzieć wspólnie w imieniu naszego ministerstwa i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, bo temat co do kompetencji jest podzielony. Przypominam, że ta pomoc doraźna w postaci zasiłków do 6 tys. została przekazana wszędzie w trybie pilnym, a jednocześnie środki na remont budynków, lokali mieszkalnych - do 200 tys., a na budynki inwentarskie - do 100 tys. zł. To nie są odszkodowania, ale pomoc dla osób najbardziej potrzebujących, żeby mogły przetrwać ten pierwszy moment po podtopieniach i zalewaniach. Jednocześnie chciałam wskazać, że na dzień 15 lipca 2020 r. z budżetu państwa przekazano na pomoc dla ponad 1940 rodzin, osób poszkodowanych łącznie prawie 17 mln. Jeżeli chodzi o jednostki samorządu terytorialnego, te straty są aktualnie szacowane, szczególnie w obrębie infrastruktury komunalnej. Po zgłoszeniu strat do wojewodów szacunki te będą podlegać weryfikacji i następnie na podstawie tych wniosków środki zostaną przekazane. Jeżeli chodzi o infrastrukturę będącą w kompetencjach Wód Polskich, straty też są aktualnie szacowane. Przypominam, że to są duże budowle hydrotechniczne, więc jeszcze chwilę potrzebujemy, żeby oszacować końcową kwotę tych strat.

Jednocześnie pozwolę sobie wspomnieć, co się udało zrobić przez te ostatnie lata, bo to są historyczne kwoty i historyczne działania. 2018 r. - w ramach kompetencji Wód Polskich wykonano łącznie 3217 zadań, w tym na wałach przeciwpowodziowych na długości prawie 5 tys. km. W 2019 r. to jest łącznie 4561 zadań, same wały przeciwpowodziowe - długość 8300.

Jednocześnie w tym roku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w ramach programu planowanych inwestycji w gospodarce wodnej zamierza prowadzić działalność inwestycyjną na 250 zadaniach inwestycyjnych, czyli tam to były zadania utrzymaniowe, to są zadania inwestycyjne, na łączną kwotę prawie miliard 700, działania przeciwpowodziowe - 113 projektów, miliard 100.

Dokończyliśmy stopień wodny Malczyce, aktualnie przystępujemy do realizacji cofki, została też wykonana część hydroenergetyczna. Aktualnie projektujemy stopnie wodne w Lubiąży i Ścinawie, co też znacząco wpłynie na funkcję przeciwpowodziową. Przypominam, że w tym roku w ostatnim momencie dokonaliśmy odbioru zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny. Historię tego zbiornika w tej Izbie nieraz państwo omawiali.

Tym samym chroni województwa śląskie, opolskie, dolnośląskie skutecznie, wystarczająco, jednocześnie zapewniając nam bezpieczeństwo w przypadku zrzutów ze strony czeskiej. Zbiorniki i inne inwestycje aktualnie wykonywane to Kąty-Myscowa, Wielowieś Klasztorna, cztery zbiorniki w Kotlinie Kłodzkiej, ochrona bierna w Kotlinie Kłodzkiej, miasto Słubice, Odra graniczna, przebudowa mostów na Odrze, Nowa Sól, węzeł wodny Widawa, kompleksowy projekt ochrony przeciwpowodziowej Sandomierza, kompleksowa rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły, rzeki Serafy w Krakowie, wał rzeki Wisły od ujścia Skawinki do stopnia Kościuszko, wał pomiędzy stopniem Dąbie a portem Płaszów, port Kujawy - brama przeciwpowodziowa, Tarnobrzeg - kompleksowa ochrona przeciwpowodziowa, gmina Tarnów - również rozbudowa wałów po obu stronach. Jednocześnie jesteśmy w fazie programowania kolejnych inwestycji. W programie przeciwdziałania niedoborom wody mamy zaplanowane 94 inwestycje. Jednocześnie kończymy planowanie programu „Stop suszy” z perspektywą (Dzwonek) 2050 r. Dziękuję. Dziękuję, pani minister. Pytanie dodatkowe, pan poseł Mieczysław Kasprzak. Dziękuję, pani minister, za te odpowiedzi, ale widocznie są to działania, jeżeli chodzi o Wody Polskie, niewystarczające, dlatego że sytuacja z roku na rok się powtarza w wielu miejscowościach i dzisiaj powiedzenie tym ludziom czy samorządom, że coś będzie za rok czy za dwa, czy za nie wiadomo ile, nie rozwiązuje problemu.

Dlatego pozwolę sobie jeszcze przekazać to pismo pani minister i prosić o to, abyście naprawdę podjęli działania skuteczne, bo samorządy mają mało pieniędzy w tym roku z wielu powodów, a przede wszystkim z tego tytułu, że o 40% dochody podatkowe spadły.

Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie pośle. Pani minister, zapraszam. Nie znam takiego, który by potrafił wybudować czy wyremontować wały w ciągu tygodnia, a rozumiem, że takie oczekiwanie pana posła tutaj aktualnie padło. Trwa szacowanie strat zarówno przez samorządy, jak i przez Wody Polskie. Po otrzymaniu tych kwot przystąpimy do realizacji prac. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Posłowie Waldemar Andzel, Jarosław Krajewski, Marek Suski, Michał Jach i Adam Śnieżek z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość zadają pytanie w sprawie ataków cybernetycznych, oszustw w Internecie, kradzieży danych i wyłudzeń. Na to pytanie z przyjemnością odpowie minister cyfryzacji pan Marek Zagórski. Zapraszam pana posła Waldemara Andzela. Wysoka Izbo! Jak podaje zespół CERT Polska, który działa w strukturach NASK, Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, najczęściej występującym typem ataków cybernetycznych na terenie naszego kraju jest phishing, czyli próba kradzieży danych, tj. loginu i hasła do kont bankowych, poczty elektronicznej i portali społecznościowych.

Należy wymienić chociażby rodzaj popularnego oszustwa internetowego, czyli tzw. metody na blika, polegającego na wyłudzeniu korzyści majątkowych, w tym wyłudzeniu pilnej pożyczki pieniężnej poprzez próbę podszycia się pod właściciela konta i kontaktowanie się z jego znajomymi lub rodziną. Inne typy oszustw to blokada systemu komputerowego dla okupu czy wysyłanie wiadomości do instytucji publicznych w celu wywołania alarmu bombowego.

W związku z tym mam pytanie do ministra cyfryzacji: Ile w sumie było zgłoszeń o naruszeniu bezpieczeństwa w sieci w roku 2019? Jaka jest liczba takich zgłoszeń w roku bieżącym?

Dziękuję serdecznie.

Rzeczywiście jest tak, że ten rok między innymi czy może przede wszystkim wskutek pandemii i zwiększonego wykorzystywania sieci jest wyjątkowy. Tak jak pan poseł powiedział, odnotowujemy zwiększoną liczbę incydentów.

Są to CSIRT NASK, odpowiadający w dużym uproszczeniu za sferę cywilną, CSIRT GOV w ABW, odpowiadający za domeny, systemy administracji rządowej, i CSIRT w Ministerstwie Obrony Narodowej, odpowiadający za sferę wojskową. Tu trzeba odróżnić: nie każde zgłoszenie jest incydentem. Te zgłoszenia podlegają analizie i w wyniku tej analizy 6484 zgłoszenia uznano za incydenty, z czego 4086 zostało zakwalifikowanych jako oszustwa komputerowe.

Trzeba powiedzieć, że tego typu ataków było 3500, przy czym te dane dotyczyły, podkreślam, 2019 r.

I to jest oczywiste, że ta aktywność w sieci obywateli, podmiotów powoduje, że jest większe zainteresowanie, większa aktywność przestępców, i widać to właśnie po tych statystykach. Jednocześnie należy podkreślić, że to, co jest pozytywne z tej strony, to większa świadomość użytkowników, bo ta większa liczba zgłoszeń jest związana z tym, że jest większa świadomość tego, w jaki sposób postępować z incydentami, z takimi przypadkami, których celem jest tak naprawdę oszustwo i wyłudzenie. Warto też powiedzieć, że w roku 2020 mieliśmy 20 incydentów poważnych. Tutaj należy zauważyć, że to jest duży wzrost w stosunku do roku poprzedniego, dlatego że w całym roku 2019 incydentów poważnych odnotowano tylko 9. Jeśli chodzi o to, jakie grupy są najbardziej narażone na ataki, to przede wszystkim chodzi o dzieci i młodzież do 18. roku życia, dlatego że one najwięcej czasu spędzają w sieci i w związku z tym są najbardziej narażone na ataki. W ogóle prowadzimy specjalne kampanie adresowane do dzieci.

Dziękuję bardzo.

Panie Ministrze! Mam pytanie dodatkowe odnośnie do fałszywych sklepów internetowych. W związku ze stanem epidemii wielu naszych rodaków zaczęło korzystać ze sklepów internetowych. Czy Ministerstwo Cyfryzacji i jednostki mu podległe odnotowały wzrost incydentów dotyczących fałszywych sklepów internetowych?

Panie ministrze, proszę. Rzeczywiście, jak już powiedziałem, największym, najbardziej powszechnym zjawiskiem jest phishing i on się przejawia m.in. tym, że to podszywanie się pod innego użytkownika jest często podszywaniem się także pod sklepy internetowe. Też warto powiedzieć, że to zjawisko, próba wyłudzeń różnego rodzaju - bo sklepy internetowe są jedną z kategorii, trzeba na to zwrócić uwagę, to zjawisko obserwowaliśmy już od samego początku pojawienia się pandemii - miało bardzo różny wymiar.

Aktualnie w rejestrze jest 2899 domen, które zostały w tym trybie zgłoszone przez operatorów, zgłoszone przez użytkowników. Następnie one przede wszystkim są blokowane, ale także informacja o tych stronach jest przekazywana organom ścigania, z którymi na bieżąco współpracują zarówno operatorzy telekomunikacyjni, jak i UKE, Ministerstwo Cyfryzacji i NASK. To, co jest istotne i co trzeba podkreślić: ten rejestr jest stworzony tylko na czas stanów nadzwyczajnych, epidemii. Każde zgłoszenie podejrzanej strony jest weryfikowane przez co najmniej dwie osoby, które się tym zajmują w CERT Polska, po to żeby uniknąć pomyłek.

Dziękuję bardzo, panie ministrze. Posłowie Michał Szczerba, Dariusz Joński i Aleksander Miszalski z Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska zdecydowali się na zadanie pytania w sprawie nieprawidłowości przy podpisywaniu i realizacji umowy na zakup 1241 respiratorów. Z pytaniem tym postara się dać sobie radę podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia pan minister Janusz Cieszyński. Zapraszam pana posła Michała Szczerbę. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Sprawa, o którą dzisiaj będziemy pytać z panem posłem Jońskim, bulwersuje opinię publiczną. Jak to jest możliwe, że byli przedsiębiorcy, którzy trafili w krąg kontrahentów Ministerstwa Zdrowia, którzy wprost chcieli zarobić na pandemii, potraktowali pandemię komercyjnie, jako okazję do zarobienia, zdobycia żyły złota? Szanowni Państwo! W ustawie tzw. tarczy 2.0 znieśliście odpowiedzialność ministrów PiS za przekroczenie uprawnień, za wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym czy naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ale, Wysoka Izbo, nie ma i nie będzie naszej zgody na to, żeby nie zajmować się sprawami, które bulwersują. Wzięto w zastaw życie i zdrowie Polek i Polaków. Zamówiono 1241 respiratorów w spółce, która zajmowała się wcześniej handlowaniem bronią. Spółce, która w ostatnich latach nie miała praktycznie żadnych obrotów, jeśli chodzi o działalność gospodarczą. Szanowni Państwo! Chcemy zadać konkretne pytania. Ile respiratorów i jakiego rodzaju odebrano protokolarnie zgodnie z umową ramową i kiedy? Ile respiratorów znajduje się w składnicach Agencji Rezerw Materiałowych i kiedy zostały dostarczone? Które ze służb weryfikowały wiarygodność kontrahenta i kiedy? Jaka część z przedpłaty wypłaconej w dniu 14 kwietnia 2020 r. została zwrócona na rachunek resortu i w jakich terminach? Ile jeszcze nie zostało zwróconych pieniędzy? Jakie kary umowne zgodnie z umową naliczył resort wobec kontrahenta i jaką kwotę udało się wyegzekwować? I kiedy odstąpiono wreszcie od umowy? Liczymy, panie ministrze, na konkretne odpowiedzi. Chcemy powiedzieć, że ta sprawa będzie dalej wyjaśniania, będzie wyjaśniana, mam nadzieję, kiedyś w ramach komisji śledczej. Dzisiaj oczekujemy konkretnych odpowiedzi przed Wysoką Izbą. Dziękuję serdecznie. Zapraszam pana ministra.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Zacznę moją odpowiedź od odczytania państwu fragmentu pisma, które wpłynęło 13 marca do Ministerstwa Zdrowia. To jest pismo skierowane do pana ministra Łukasza Szumowskiego. Szanowny Panie Ministrze! Na podstawie art. 16 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja o wykonywaniu mandatu posła i senatora wobec postępującej w dynamicznym tempie liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2 wnosimy o pilne dokonanie zakupu respiratorów niezbędnych w leczeniu choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2. To jest, szanowni państwo, pismo z marca, kiedy państwo jeszcze byli gotowi w uczciwy sposób współpracować z rządem przy zwalczaniu epidemii i kiedy państwo sami widzieli, że jest potrzeba dokonywania zakupów. Później sytuacja się zmieniła, ponieważ widzieliście, że wasz kandydat w wyborach prezydenckich nie ma szans, co się zresztą potwierdziło w ostatecznym wyniku, i postanowiliście zaatakować. Zgodnie ze starą polityczną zasadą zaatakowaliście tam, gdzie byliśmy najmocniejsi, czyli tam, gdzie.

I dlatego zaczęło się od wysłania forpoczty w postaci pana Nitrasa, który wtargnął na briefing do Ministerstwa Zdrowia. No a później przyszli panowie, przyszliście panowie i mówiąc opinii publicznej, że domagacie się wyjaśnień, tak naprawdę robiliście polityczne show. Każdy to widział. To, co was najbardziej interesowało, to zrobienie briefingu. Najlepszym przykładem jest sytuacja, kiedy otrzymali panowie potwierdzenia przelewów środków, które wróciły na konto Ministerstwa Zdrowia. Zgadnijcie państwo, co zrobili panowie posłowie po tym, kiedy otrzymali tę informację, której tak bardzo się domagali. Zrobili briefing pod siedzibą Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a o faktach nie powiedzieli nic. Ale o faktach powiem ja. Powiem to po raz kolejny, ponieważ od samego początku transparentnie i uczciwie rozliczamy się z całej tej sprawy. Pytacie państwo, ile respiratorów. 200 sztuk, 50 firmy Dräger, 150 firmy Mekics, odebranych 30 czerwca tego roku. Ile środków wróciło na konto Ministerstwa Zdrowia? Do tej pory wróciło już ponad 14 mln euro. Mamy informację o tym, że kolejne środki też do nas wrócą.

Za opóźnienie nałożyliśmy odpowiednie odsetki. Od samego początku, szanowni państwo, ta umowa jest realizowana w całości, w pełni w interesie Skarbu Państwa. Takie są fakty na temat tej transakcji i żadne kolejne występy panów posłów tego nie przykryją. Dziękuję serdecznie. Pytanie dodatkowe zada pan poseł Dariusz Joński, Koalicja Obywatelska. Dziękuje. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szkoda, że to tylko 1 minuta, ale postaram się krótko. Najpierw był parasol ochronny, czyli ustawa, która mówiła o bezkarności tych, którzy robili zamówienia.

Chodzi o brak odpowiedzialności za to, że tych respiratorów nie ma. W kwietniu zamówiliście u handlarza bronią, bo myśleliście, że on to sprzeda. Było wiadomo, że nie ma żadnego doświadczenia. I to pytanie chciałbym zadać panu premierowi Morawieckiemu. Panie ministrze, zapraszam.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Wobec powyższego bardzo mi przykro, ale muszę pozostawić pana pytanie bez odpowiedzi. Pytał mnie pan, czy prawdą jest to, że brakuje 90 mln. Nie, proszę pana, to jest kłamstwo, kolejne pana kłamstwo. Proszę państwa, posłowie Krzysztof Gawkowski, Tadeusz Tomaszewski, Karolina Pawliczak, Katarzyna Kretkowska, Anita Sowińska, Wiesław Szczepański i Marcelina Zawisza z klubu Lewica postanowili zadać pytanie w sprawie przeprowadzenia zwolnień grupowych i rozpoczęcia procedury konsultacji w sprawie zwolnień grupowych w PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów SA oraz PAK Górnictwo sp. z o.o. - spółkach zależnych od grupy kapitałowej Zespół Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin SA. Pytanie to zostało skierowane na ręce prezesa Rady Ministrów, a odpowie na to pytanie sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pan minister Stanisław Szwed. Bardzo proszę pana posła Tadeusza Tomaszewskiego z klubu parlamentarnego Lewica. Proszę bardzo. Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Szanowny Panie Ministrze! 1 stycznia przestała funkcjonować Elektrownia Adamów, a w maju 2020 r. ogłoszono decyzję o zaprzestaniu dalszej eksploatacji węgla w odkrywce Adamów na terenie powiatu tureckiego.

W wyniku decyzji wspomnianych spółek rozpoczęła się procedura zbiorowych zwolnień.

W tej chwili po konsultacjach ze związkami zawodowymi będzie to 187 górników na terenie jednego powiatu, powiatu tureckiego. To wszystko powoduje, że trzeba działań osłonowych ze strony państwa. Nie wystarczą instrumenty znane na rynku pracy, bo w tej chwili pracodawca wobec zwalnianych górników zastosował tylko i wyłącznie procedury wynikające ze zwolnień grupowych, czyli odprawy jedno-, dwu- i trzymiesięczne. Dlatego też domagają się, aby zastosować wobec nich takie systemy osłonowe jak urlopy górnicze, emerytury pomostowe, zasiłki socjalne, jednorazowe odprawy, udzielanie pożyczek na preferencyjnych zasadach w celu podjęcia działalności gospodarczej. Uważają, że mają prawo, zgodnie z konstytucją, być traktowani na tożsamych zasadach jak górnicy z branży węgla kamiennego. Dlatego też w imieniu (Dzwonek) tychże górników, ale także działaczy związkowych uprzejmie proszę rząd o podjęcie stosownych działań zapobiegających katastrofie wynikającej z zakończenia działalności przemysłu wydobywczego na terenie powiatu tureckiego. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. pana ministra Stanisława Szweda. Panie Marszałku! Panie Pośle!

Jeśli chodzi o zwolnienia, 18 maja zarząd zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników zgłosił zamiar zwolnień grupowych. Zgodnie z procedurą zgłosił to do związków zawodowych. Trwają w tym zakresie negocjacje.

Oczywiście na to też nakłada się fakt taki, tu przechodzę do pytania dotyczącego programu osłonowego, że dzisiaj dotyczy to jednak jeszcze dosyć wąskiej grupy pracowników, jeśli chodzi o zwolnienia. Mamy też, jeśli chodzi o Wielkopolskę, dobrą sytuację na rynku pracy, bo województwo wielkopolskie zawsze szczyci się tym, że ma najniższą stopę bezrobocia, choć ten region, o którym mówimy, w tym województwie jest tym regionem, gdzie to bezrobocie jest wyższe.

W tym zakresie nie mamy jakiegoś specjalnego instrumentu, tylko korzystamy z tych instrumentów, które są w powiatowych urzędach pracy, zarówno w Turku, jak i w Koninie.

I takie środki, oczywiście jeżeli będzie takie zapotrzebowanie, uruchomimy. Dzisiaj te środki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w tych urzędach są uruchamiane, one funkcjonują, tak że można też z tych informacji skorzystać. To jest kwestia wystąpień, które wpłynęły do pana premiera Sasina. Szansą na rozwiązanie problemów PAK, Kopalni Węgla Brunatnego Adamów jest skorzystanie ze wsparcia oferowanego w ramach Platformy Regionów Górniczych w Procesie Transformacji, której celem jest zbieranie projektów mogących wspomóc transformację regionów górniczych. Komisja Europejska w 2018 r. wytypowała 41 regionów górniczych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W Polsce wskazano sześć takich obszarów. Zakwalifikowanie przez Komisję Europejską danego regionu jako region górniczy otwiera możliwość przystąpienia do takiego programu.

Pytanie dodatkowe zada pan poseł Tomaszewski Tadeusz. Zapraszam. Panie Marszałku! Szanowny Panie Ministrze! Powiedział pan tylko i wyłącznie o instrumentach rynku pracy. Niestety sytuacja w związku z likwidacją sektora paliwowo-energetycznego wymaga szerszych działań osłonowych ze strony rządu. Tak, rzeczywiście wczoraj pan premier Sasin, odpowiadając na moją interpelację, powiedział m.in.: jednakże na chwilę obecną nie ma programu osłon socjalnych dla pracowników sektora węgla brunatnego.

Zwolnienia dzieją się dzisiaj, dzisiaj ludzie potrzebują nowych miejsc pracy.

To kolejne zwolnienia grupowe w tej części Wielkopolski (Dzwonek), a więc te instrumenty mogą okazać się za małe.

Dziękuję. Panie ministrze, zapraszam. Panie Pośle! Tutaj oczywiście można było podać też informacje dotyczące funkcjonowania tarczy antykryzysowej, tarczy finansowej, która przecież też mocno wspiera ochronę miejsc pracy. Dotyczy to również województwa wielkopolskiego i tego regionu, o którym mówimy.

Dziękuję serdecznie. Posłowie Barbara Bartuś, Joanna Borowiak i Lidia Burzyńska z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość postanowiły zadać pytanie w sprawie działań podjętych przez żołnierzy WOT w czasie epidemii koronawirusa w zakresie niesienia pomocy służbom, m.in. medycznym i sanitarnym, oraz udzielania wsparcia obywatelom. Na to pytanie odpowie minister obrony narodowej pan Mariusz Błaszczak. Zapraszam panią poseł Barbarę Bartuś. Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Wojska Obrony Terytorialnej utworzone 1 stycznia 2017 r. na mocy ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z 16 listopada stanowią znaczne wzmocnienie Wojska Polskiego. Stoją na posterunku zawsze tam, gdzie są potrzebne. Cieszę się bardzo, że wojska te są doceniane też przez całe ministerstwo i że dzisiaj osobiście na nasze pytanie w tym temacie odpowiada minister Mariusz Błaszczak, bo to jest minister stojący na czele resortu, który dba o bezpieczeństwo naszego kraju, naszej ojczyzny, i to w każdym zakresie. Wojska Obrony Terytorialnej są też wszędzie tam, gdzie ludzie potrzebują pomocy.

Pamiętamy początek marca, ten strach i pamiętamy Wojska Obrony Terytorialnej, które były wszędzie tam, gdzie była potrzebna pomoc. I dlatego chciałabym zapytać pana ministra: Jaka liczba żołnierzy brała udział w działaniach wspierających walkę z koronawirusem w kraju i jak to wyglądało w poszczególnych regionach, w poszczególnych województwach? Jakie działania wykonywali żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej w trakcie walki z epidemią? Czy ta pomoc została też doceniona przez Polaków? Dziękuję bardzo. Witam serdecznie pana ministra Mariusza Błaszczaka i zapraszam na mównicę. Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Bardzo dziękuję za to pytanie zgłoszone przez panie posłanki. Chciałbym podkreślić bardzo ważną rolę Wojsk Obrony Terytorialnej w sytuacjach kryzysowych. Chciałbym podkreślić, że w moim głębokim przekonaniu, ale nie tylko moim, bo również ludzi, z którymi miałem sposobność rozmawiać, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej sprawdzili się. Są zawsze gotowi, są zawsze blisko. Nieśli oni pomoc poszkodowanym zarówno w czasie epidemii, jak i w czasie podtopień. Choćby ostatnio, 2 tygodnie temu podczas fali podtopień na południu Polski, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej byli na miejscu. Wysoka Izbo! Epidemia koronawirusa była jednym z największych zagrożeń ostatnich dekad. Jednak przyniosła ona ze sobą także jeden pozytyw. Już nikt w Polsce nie może mieć wątpliwości co do przydatności Wojsk Obrony Terytorialnej. Determinację, upór i zaangażowanie osób służących w WOT mogliśmy obserwować każdego dnia walki z pandemią. Swoje wystąpienie chcę rozpocząć od podziękowań za tytaniczną pracę, którą żołnierze wykonywali i wciąż wykonują. Każdy z nas, parlamentarzystów, powinien pochylić czoło przed żołnierzami w oliwkowych beretach. To nasza powinność. Moje wystąpienie dotyczy Wojsk Obrony Terytorialnej, ale nie wolno nam zapominać, że podziękowania należą się także wojskom operacyjnym oraz wojskowym medykom. Wysoki Sejmie! Bilans wsparcia WOT podczas epidemii robi wrażenie i całkowicie potwierdza potrzebę powołania tej formacji. To pomoc udzielana setkom szpitali, domów pomocy społecznej, placówek oświatowych oraz organizacji społecznych. Już w marcu podpisałem decyzję, na mocy której żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej i Żandarmerii Wojskowej wspierali Policję podczas patrolowania ulic i kontrolowania przestrzegania kwarantanny. Pandemia wyjątkowo silnie uderzyła w domy pomocy społecznej, których pensjonariusze są szczególnie narażeni na infekcję.

Żołnierze udzielali wsparcia w ewakuacji, w przywracaniu zdolności do funkcjonowania domów pomocy społecznej. Transportowali pensjonariuszy placówek, m.in. w Drzewicy czy Koleczkowie, ewakuowali domy pomocy społecznej w Pleszewie, Czernichowie i Kaliszu. WOT udzieliły wsparcia w ponad 536 domach pomocy społecznej, a żołnierze pozostawali w kontakcie z dyrekcją wszystkich ponad 800 placówek w Polsce. Wojska Obrony Terytorialnej otoczyły opieką ponad 3 tys. osób starszych, kombatantów, rodzin medyków i osób samotnych. Przetransportowali ponad 40 tys. t żywności i ponad 260 tys. paczek ze środkami ochrony osobistej do potrzebujących oraz zrealizowali ponad 700 transportów z ponad 7,5 tys. t towarów dostarczonych do 2 tys. miejsc dystrybucji. Pomoc Wojsk Obrony Terytorialnej w diagnozowaniu pacjentów była nieoceniona. W miejscach trudno dostępnych i w sytuacjach, gdzie liczy się przede wszystkim szybkość działania, z pomocą przychodziły mobilne punkty do pobierania próbek, czyli test and go, które były obsługiwane przez żołnierzy. Część z nich ciągle działa. Z inicjatywy terytorialsów powstała także bezpłatna infolinia z pomocą psychologiczną, która udzielała wsparcia osobom w kryzysie. Z czasem przerodziła się ona w bezpośrednią pomoc dla rodziców, którzy musieli organizować swoim dzieciom zdalną naukę. Obecnie WOT pomaga organizatorom kolonii i obozów harcerskich w przygotowaniu bezpiecznych wakacji. Wysoka Izbo! Skala zaangażowania żołnierzy WOT tym bardziej robi wrażenie, że są to ochotnicy, najczęściej posiadający również inne zobowiązania zawodowe. Dziwią więc głosy wielu przedstawicieli opozycji, którzy wciąż powtarzają o konieczności reformowania WOT lub nawet likwidacji. Podkreślam: nie pozwolę ruszyć Wojsk Obrony Terytorialnej. Nie pozwolę zdusić zapału tych [[Oklaski]] patriotyczne nastawionych wspaniałych ludzi, bez których walka z epidemią (Dzwonek) nie byłaby możliwa. Dziękuję serdecznie, panie ministrze. Pytanie dodatkowe zada pani poseł Joanna Borowiak. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Dziękuję serdecznie za tę informację, której pan udzielił. Skala zaangażowania ochotników, żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej nie tylko w służbę, ale także w pomoc niesioną ludziom, jest naprawdę ogromna. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej są doceniani przez społeczeństwo, ale niestety nie są doceniani przez wszystkich parlamentarzystów, szczególnie przychodzą mi na myśl sformułowania używane przez posłów Platformy Obywatelskiej, którzy próbowali w ostatnim czasie zdeprecjonować i ośmieszyć żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Padały takie sformułowania jak „bieganie z drewnianymi pukawkami” czy też oskarżenia, że nie mają ćwiczeń, nie potrafią strzelać itd. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej są tym zbulwersowani, bo bardzo wiele takich głosów otrzymałam. Na ręce pana ministra składam serdeczne podziękowania dla nich za ofiarność w pełnieniu służby, za ofiarność w niesieniu pomocy, szczególnie pomocy seniorom. I jeszcze pytanie, panie ministrze. Jak na chwilę obecną wygląda sytuacja w zakresie liczebności Wojsk Obrony Terytorialnej i ich rozmieszczenia w Polsce? Dziękuję. Dziękuję, pani poseł. Panie ministrze, zapraszam serdecznie. Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Chciałem podkreślić, że Wojska Obrony Terytorialnej sprawdziły się, że Wojska Obrony Terytorialnej, mam nadzieję, mam pewność, na stałe wpisały się w krajobraz funkcjonowania służb w sytuacjach kryzysowych. Słyszałem od bardzo wielu osób słowa podziękowania za to, że żołnierze WOT-u byli na służbie, byli o czasie, że pomagali. Chciałbym też - podkreślam - podziękować panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie, który wspierał - i deklaruje dalsze pełne jego wsparcie - rozwój najmłodszego rodzaju Sił Zbrojnych. To jest niezwykle istotne, żeby Wojska Obrony Terytorialnej się rozwijały. Podam kilka liczb mówiących o tym, że ten proces następuje i następuje dynamicznie. Otóż na koniec 2017 r. Wojska Obrony Terytorialnej liczyły 7600 żołnierzy, na koniec ubiegłego roku było to 24 300 żołnierzy. Przed chwilą rozmawiałem z panem pułkownikiem - w ciągu miesiąca, zaledwie w ciągu miesiąca 1100 żołnierzy przystąpiło do Wojsk Obrony Terytorialnej. To świadczy [[Oklaski]] o dużym zaangażowaniu, dużym poczuciu patriotyzmu, ale też chęci służenia innym ze strony ludzi, którzy poświęcają przecież część swojego wolnego czasu, żeby właśnie służyć innym. Rozwija się liczebnie struktura Wojsk Obrony Terytorialnej, jest to proces, który przebiega bez zakłóceń. I jeszcze kilka informacji ogólnych dotyczących zaangażowania w walkę z koronawirusem. Otóż ogólna liczba zaangażowanego personelu WOT w tym czasie to 20 347 osób. Ogólna liczba wspartych podmiotów medycznych - 632, w tym 496 szpitali, 118 placówek medycznych, 18 izb pielęgniarskich. Ogólna liczba transportów żywności do ośrodków pomocy społecznej oraz organizacji non profit z banków żywności to 5603. Może jeszcze ogólna liczba honorowych dawców krwi - 6232, może jeszcze ogólna ilość żywności w tonach dostarczonej do ośrodków pomocy społecznej - 48 tys. t. Wysoki Sejmie! W czasie epidemii terytorialsi byli wszędzie tam, gdzie ich potrzebowaliśmy. Jeszcze raz chcę stanowczo podkreślić: likwidacja WOT to krzywdzenie państwa i działanie na szkodę naszej ojczyzny. Nie dopuścimy do tego. Dziękuję serdecznie. Przechodzimy do pytania pań posłanek Iwony Hartwich i Ewy Kołodziej z Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska. Pytanie będzie dotyczyło osób z niepełnosprawnością po 18. roku życia, które nie zostały ujęte w ustawie o Polskim Bonie Turystycznym. Na to pytanie będzie odpowiadał sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju pan minister Andrzej Gut-Mostowy. Bardzo proszę panią posłankę Iwonę Hartwich. Twoja jest mównica. Szanowny panie Marszałku! Wysoka Izbo! Rządzie PiS! Prezydencie Andrzeju Duda! Osoby z niepełnosprawnością zostały przez was oszukane. Kolejny raz zostały oszukane.

Ustawa tzw. 520 zł, głoszona i promowana przez panie minister Rafalską i Kopcińską, okazała się zwykłym oszustwem. Żadna z osób z niepełnosprawnościami do dzisiaj nie zaoszczędziła nawet złotówki. Przez cały okres waszych rządów oszczędzacie na osobach z niepełnosprawnościami. Boicie się obliczyć dla nich minimum socjalne. Doskonale wiecie, że ta głodowa renta socjalna, która jest głęboko niewystarczająca, oznacza brak szans na godne życie, na rehabilitację, na leczenie. Podczas pandemii znów okradliście najsłabszych, znów okradliście osoby z niepełnosprawnościami.

Czy zabrakło wam środków, a może chęci? Bo na pewno zabrakło wam empatii. Przestańcie dyskryminować osoby niepełnosprawne, przestańcie dzielić. Są normy przyzwoitości. Moje pytanie. Dlaczego rząd PiS nie ujął w ustawie o Polskim Bonie Turystycznym osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji po 18. roku życia, pobierających świadczenie uzupełniające w kwocie 500 zł? Dziękuję, pani poseł. Bardzo proszę pana ministra Andrzeja Gut-Mostowego. Witam serdecznie. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowne Posłanki! Polski Bon Turystyczny jako projekt pana prezydenta jest projektem, który łączy elementy polityki społecznej. czyli każde dziecko uprawnione do 500+ otrzyma świadczenie w wysokości 500 zł, przy czym dodatkowe środki zostaną także przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, a także dla osób znajdujących się w tzw. koordynacji świadczeń europejskich. Zazwyczaj są to rodziny, w których jeden rodzic pracuje za granicą. Z programu będzie mogło skorzystać ponad 6 mln dzieci. Według danych i tendencji w rodzinach można oszacować liczbę dzieci urodzonych w latach 2020 i 2021 na ok. 740 tys. Polskie rodziny otrzymają 500 zł na każde dziecko niezależnie od tego, jakie mają zarobki, tak jak w przypadku programu 500+. Osobom wychowującym dzieci z niepełnosprawnością będzie przysługiwało dodatkowe świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł na każde dziecko, czyli łącznie 1 tys. zł.

Ustawa obejmie dzieci legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym albo znacznym, czyli dotyczy to wszystkich rodzajów niepełnosprawności.

Co istotne, jest to projekt wyjątkowy na skalę europejską. Nie ma takich projektów, które by w taki sposób łączyły elementy polityki społecznej i polityki gospodarczej, stymulując turystykę, która tak mocno została dotknięta przez epidemię COVID.

Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Pytanie dodatkowe, pani posłanka Iwona Hartwich. Wysoka Izbo!

Obiecywał to w trakcie protestu. Tak samo jak osoby z niepełnosprawnościami państwo, nie dając im szansy na wypoczynek, bo uważacie, że im się nie należy, oszukaliście emerytów i rencistów. Obiecaliście im bon turystyczny w kwocie 1000 zł. Tuż po wyborach pamięć straciliście. Prezydent i rząd muszą wywiązywać się ze swoich obietnic. I jednak uważam, że te opowieści z mchu i paproci to tak naprawdę wychodzą (Dzwonek) panu Mateuszowi Morawieckiemu. Czy waszym zdaniem również tej grupie, emerytom i rencistom, nie należy się pomoc? Dziękuję serdecznie. Zapraszamy ponownie pana ministra z prośbą o odpowiedź, dlaczego tak się wydarzyło. Wysoka Izbo! Szanowne Posłanki! Polski Bon Turystyczny jest skierowany do ok. 6 mln dzieci.

Co też jest istotne, jako że Ministerstwo Rozwoju współpracowało z Kancelarią Prezydenta i służyło swoją wiedzą i swoim doświadczeniem, bardzo ważne było - aby ten projekt został uruchomiony już w lipcu lub w sierpniu, czyli w przeciągu 2–3 tygodni - aby baza tych beneficjentów bonu turystycznego była jasno sprecyzowana i można było ją szybko utworzyć, aby można było już w sierpniu wypłacać środki w ramach Polskiego Bonu Turystycznego, bo branża turystyczna na to czeka.

Dziękuję serdecznie. Posłowie Marek Polak i Leonard Krasulski z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość zadają pytanie w sprawie inwestycji infrastrukturalnych w dobie kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa. Na to pytanie będzie odpowiadał sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury pan minister Rafał Weber, którego serdecznie witamy. Dziękuję bardzo. Szanowny Panie Marszałku! Szanowny Panie Ministrze! Kryzys gospodarczy wywołany pandemią koronawirusa wybuchł w Polsce w czasie, gdy na terenie całego kraju trwa realizacja dużych projektów infrastrukturalnych, z których najważniejsze to budowa przekopu Mierzei Wiślanej, a także przygotowania do budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Warto również wspomnieć, że na terenie całej Polski trwa realizacja innych licznych zadań drogowych, jak również kosztownych inwestycji kolejowych. Pojawiły się zatem obawy, że w obecnej sytuacji realizacja tych inwestycji może być zagrożona. Takie opinie były też podnoszone w wypowiedziach niektórych opozycyjnych kandydatów na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w trakcie minionej kampanii wyborczej, którzy wprost nawoływali do zawieszenia tych inwestycji. Dlatego chciałbym zapytać, czy pandemia koronawirusa rzeczywiście ma negatywny wpływ zarówno na terminowość, jak i celową realizację tych zadań. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Zapraszam pana ministra.

Wysoka Izbo! Szanowni Państwo! Chyba każdy z nas miał obawy na początku marca, gdy epidemia koronawirusa na świecie, w Europie bardzo mocno dała się we znaki. Wtedy również Ministerstwo Infrastruktury i ci, którzy prowadzą w naszym imieniu inwestycje i drogowe, i kolejowe, mieli obawy, czy nie wpłynie to na terminowość prac realizacyjnych, na terminowość prac budowlanych. I od samego początku zarówno pan premier Mateusz Morawiecki, jak i pan minister Andrzej Adamczyk tak tworzyli, tak konstruowali obszar prawny, aby nie tylko utrzymać wszystkie inwestycje drogowe, kolejowe, które są prowadzone, ale również ten stan prawny poprawić, ulepszyć i przeznaczyć większe środki finansowe na inwestycje publiczne. I po 5 miesiącach od początku epidemii koronawirusa możemy powiedzieć z czystym sumieniem, z ręką na sercu, że epidemia nie wpłynęła na terminowość prac realizacyjnych zarówno drogowych, jak i kolejowych. Jest to wynik doskonałej współpracy całej branży budowlanej. Jest to wynik, tak jak powiedziałem, rozsądnych, roztropnych i trafnych decyzji rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego, pana ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka. Jest to wynik działań, które prowadzili i prowadzą nadal zamawiający publiczni, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a także spółki kolejowe PKP PLK i PKP SA. Koronawirus polskich budów nie zatrzymał.

Wszystkie programy, które były realizowane na początku tego roku, są realizowane również po tym okresie 5 miesięcy trwania epidemii, również „Program budowy dróg krajowych na lata 2014-2023”, a w ramach tego programu w tej chwili prawie 100 zadań inwestycyjnych: budowa ciągów autostradowych, budowa ciągów dróg ekspresowych, budowa obwodnic. To wszystko jest prowadzone, to wszystko jest realizowane. Tak samo zresztą jak inne inwestycje drogowe na sieci: modernizacja dróg już istniejących, dostosowanie do 11,5 t nacisku na oś, zadania polegające na poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, modernizacja wiaduktów, mostów. To łącznie blisko 600 tytułów inwestycyjnych, które są w tej chwili realizowane na drogach krajowych. Trzeba również dodać do tych inwestycji niezahamowane inwestycje samorządowe i finansowanie inwestycji samorządowych, Fundusz Dróg Samorządowych. Pan premier 15 kwietnia zatwierdził listę zadań i gminnych, i powiatowych, blisko 2300 tytułów inwestycyjnych, które są też realizowane przez gminy i przez powiaty. A w poprzednim tygodniu wojewodowie ogłosili nabory na rok 2021, tak że konsekwentnie i systematycznie Fundusz Dróg Samorządowych jest prowadzony, jest realizowany. Finansowanie przez rząd Prawa i Sprawiedliwości jest zapewnione, zresztą tak samo jak finansowanie innych mechanizmów wspierających budownictwo drogowe lokalne. Rezerwa subwencji ogólnej - ona też przy współpracy z Ministerstwem Finansów została zatwierdzona. 110 tytułów inwestycyjnych, 110 zadań drogowych w województwach i w miastach na prawach powiatu, a także w polskich powiatach dzięki temu wsparciu jest w roku 2020 realizowanych. Tutaj mamy 230 tytułów inwestycyjnych. Jest program inwestycji dworcowych realizowany przez PKP SA. Tutaj mamy 189 tytułów inwestycyjnych. Jest program „Kolej+”, który jest dedykowany samorządowcom, by odtworzyć te linie o znaczeniu regionalnym. Nabór trwa. Widzimy duże zainteresowanie samorządów. Mamy nadzieję, że przerodzi się to w złożone wnioski, tak aby te bardzo istotne połączenia kolejowe, istotne z punktu widzenia regionalnego, były realizowane. Tak że, szanowni państwo, nie tylko inwestycje nie zostały wstrzymane, ale również dzięki, tak jak powiedziałem, dobrym, rozsądnym, roztropnym decyzjom i prawnym, i finansowym te inwestycje są prowadzone. A najdobitniejszym przykładem tego, że chcemy jak największe środki inwestować w inwestycje publiczne, jest zmiana programu budowy dróg krajowych i poszerzenie limitu o kolejne 22 mld zł, tak aby zrealizować drogę ekspresową S6 na Pomorzu czy odcinek drogi ekspresowej S10 od Bydgoszczy do Torunia. I CPK jest w fazie przygotowawczej, i inwestycje polegające na przekopie Mierzei Wiślanej, chociaż jest to prowadzone przez inny resort, również przebiega zgodnie z planem, zgodnie z harmonogramem. Tak że jeszcze raz gorąco dziękuję wszystkim tym, którzy przez ostatnie 5 miesięcy solidnie pracowali na to, i pracują nadal, aby inwestycje drogowe, kolejowe były realizowane zgodnie z harmonogramem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie Ministrze! Dziękując za te wyczerpujące i optymistyczne informacje, chciałbym jeszcze w kilku słowach nawiązać do licznych wypowiedzi pana ministra Andrzeja Adamczyka, który stanowczo zapewnia, że wszystkie zaplanowane inwestycje zarówno drogowe, jak i kolejowe, pomimo pandemii koronawirusa, będą kontynuowane, i zapewnia też, że realizacja tych zadań z jednej strony pozwala na organizowanie pracy w sposób bezpieczny dla zdrowia pracowników na placu budowy, a z drugiej strony ma trwałe i stabilne finansowanie, przy czym sprzyjająca pogoda może dać wyniki jeszcze wyższe od pierwotnie zakładanych. Ale korzystając z okazji, chciałbym pana ministra zapytać, a właściwie prosić, aby pan minister potwierdził, ewentualnie zaprzeczył: Czy te optymistyczne i dobre informacje nadal są aktualne i czy nic się nie zmieniło oraz czy nic temu nie zagraża? Dziękuję bardzo. Panie ministrze, niech pan pochwali jeszcze raz swój resort. Z przyjemnością się tego słucha. Proszę bardzo. Dlatego wykorzystam te prawie 3 minuty, aby jeszcze raz podkreślić to, że inwestycje publiczne drogowe i kolejowe nie tyle nie są wstrzymane, ile ich zakres jest poszerzany. Szanowni państwo, epidemia COVID-19 jeszcze bardziej zbliżyła resort infrastruktury i zamawiających do branży wykonawczej. Mieliśmy spotkania w interwale niemalże kilkudniowym, gdzie na bieżąco ze wszystkimi wykonawcami, tymi największymi, inwestycji drogowych i kolejowych omawialiśmy problemy, które występują na budowach i, tak jak mówię, podejmowaliśmy działania prawne zmierzające do rozwiązywania tych problemów. Szanowni państwo, to przyniosło skutek, to przyniosło efekt. Chcemy tę zbliżoną współpracę oczywiście podtrzymywać teraz. Jeszcze raz bardzo gorąco dziękuję całej branży wykonawczej, wszystkim firmom wykonawczym, podwykonawcom, organizacjom zrzeszającym tę branżę za taką bardzo ścisłą, dobrą i efektywną współpracę, licząc, że po ustabilizowaniu się sytuacji zdrowotnej ta współpraca będzie cały czas na takim samym, bardzo dobrym poziomie.

Tak jak powiedziałem, w samym epicentrum tej epidemii, czyli w kwietniu, pan premier zatwierdził listę, jeśli chodzi o Fundusz Dróg Samorządowych w roku 2020, natomiast w poprzednim tygodniu wojewodowie ogłosili nabór na rok 2021.

Dziękuję, panie pośle, za pytania, za zainteresowanie tym tematem. Szacujemy, że w branży budowlanej pracuje ok. 1,5 mln osób - to są budowlańcy, to są pracownicy firm kooperujących, dostawcy - i naprawdę finansowanie tych inwestycji nie tylko jest niezbędne do poprawy komunikacyjnej, do skracania dystansów, do poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego, ale również jest niezbędne do tego, aby podtrzymać wysoki poziom gospodarczy. I to też w trakcie epidemii zdrowotnej ma kolosalne znaczenie. Po pana słowach aż się chce ruszyć w drogę.

Na pytanie to będzie odpowiadał podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju pan minister Marek Niedużak, którego serdecznie witamy. Proszę bardzo, pytanie zada pani poseł Monika Wielichowska. Proszę. Dziękuję, panie marszałku. Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Branża kreatywna, branża artystyczna przez pandemię jest w niebywale trudnej sytuacji. Została zamrożona jako pierwsza i do dziś nie pracuje. Tysiące ludzi pozostało bez możliwości zarobkowania z dnia na dzień, z leasingami, z kredytami i z niepewną przyszłością. Bez odmrożenia tego sektora, bez odpowiedniego czasu, by podnieść branżę z kryzysu, i bez popytu na usługi branża bezpowrotnie zniknie z polskiego rynku. Mimo luzowania obostrzeń powrót do normalności w tym sektorze nie jest możliwy, ponieważ kryzys gospodarczy przełożył się na wycofanie publicznych i prywatnych inwestorów. Branża stanowi 3,5% PKB i jest istotnym elementem polskiej gospodarki, którą buduje praca techników estradowych, realizatorów dźwięku, światła, riderowców, animatorów, konstruktorów, muzyków, artystów, agentów, producentów. To ponad 300 tys. miejsc pracy. To wszyscy ci, którzy swoją profesjonalną pracą na światowej klasy sprzęcie, najczęściej leasingowanym i w kredytach, składają się na efekt końcowy każdego artystycznego wydarzenia, każdego festiwalu, koncertu, konferencji czy eventu. To branża, która wymaga indywidualnego spojrzenia i pomocy państwa, bo ten sektor nie stanie na nogi w tym roku. Czy rząd wie, że przez pandemię w tym roku nie odbędzie się 7200 imprez masowych, nie będzie tysięcy imprez biletowanych i ponad 7 tys. koncertów się nie odbędzie? Czy rząd wie, że właściciele firm technicznych z powodu braku zleceń, braku pracy nie są w stanie płacić rat leasingowych i są oddawani w ręce komorników i windykatorów jak pospolici oszuści? Co rząd zrobił do tej pory, by pochylić się nad postulatami branży? Czy rząd nawiązał dialog z Polską Izbą Techniki Estradowej lub Izbą Gospodarczą Menedżerów Artystów Polskich? To izby przedsiębiorcze branży, które od tygodni [[Dzwonek]] proszą o pomoc, informują o swoich problemach i przygotowały pakiet propozycji, które pomogłyby im przetrwać - „Otwieramy koncerty” Czy ich widać, czy ich słychać? Bo oni protestują. Które z ich postulatów zostaną uwzględnione w kolejnej tarczy? Na jakim etapie jest wypracowywanie mapy drogowej powrotu do normalnych zasad funkcjonowania branży kreatywnej, branży, panie ministrze, która bez pomocy państwa nie przetrwa? Zapraszam pana ministra. Wysoka Izbo! Pani Poseł! Mówię w imieniu ministra rozwoju, aczkolwiek oczywiście jest to pole przede wszystkim ministra kultury. Jeśli chodzi o spotkania pani premier Emilewicz z branżą rozrywkową i koncertową, to mam informacje o trzech takich spotkaniach.

Tak że jak najbardziej jesteśmy w bieżącym kontakcie z przedstawicielami tej branży i zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to branża szczególnie dotknięta trudną sytuacją. Proszę zwrócić uwagę zresztą na to, że ogniska chorób pojawiają się bardzo często przy okazji, dozwolonych oczywiście, nie wiem, ślubów, wesel, i prawdę mówiąc, obawiam się, że impreza typu koncert w jakiś sposób podobne ryzyko mogłaby rodzić. Natomiast by być troszkę bardziej specyficznym, to chciałbym zwrócić uwagę na harmonogram odmrażania tej branży. To są informacje, które mam od ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Od 6 czerwca jest możliwe prowadzenie działalności kulturalnej i rozrywkowej w pomieszczeniach, amfiteatrach oraz muszlach koncertowych przy założeniu, że mamy co drugie miejsce, rzędy są naprzemienne. Od 20 czerwca - w salach koncertowych, klubach muzycznych, halach widowiskowo-sportowych, w amfiteatrach, muszlach koncertowych przy założeniu, że mamy 50% zapełnionych miejsc na sali. Od 20 czerwca - w obiektach sportowych na wolnym powietrzu, a od 17 lipca również organizowanie wydarzeń na otwartej przestrzeni bez limitu 150 osób pod warunkiem zachowania dystansu społecznego. Z tego, co mi wiadomo, Ministerstwo Rozwoju, ministerstwo kultury wspólnie z ministrem zdrowia i głównym inspektorem sanitarnym prowadzi konsultacje na temat ewentualnej możliwości dalszego znoszenia tych ograniczeń.

Zdaję sobie sprawę, że tej pomocy nigdy nie będzie dość, prawda.

Ale tak jak mówię, w historii III RP jeszcze się nie zdarzyło, aby o ludzi współpracujących w takiej formie państwo się zatroszczyło, a zdaję sobie sprawę, że w tej branży bardzo dużo ludzi współpracuje w takiej formie. Są też inne formy pomocy, chociażby rozwiązanie dotyczące voucherów i zwrotu kwoty wpłaconej już przez klientów w ciągu 180 dni. Tak że to nie jest tak, że państwo o tej branży nie myśli. Środki pomocowe zostały tam skierowane, pewne rozwiązania pomocowe zostały przyjęte i staramy się ją odmrażać, ale to wszystko musi być w odpowiednim rygorze sanitarnym, musimy pamiętać o tym, że mamy pandemię.

już abstrahując od tej firmy, o której myślę w tej chwili, od marca - żadnego. Rozumiem całą sprawę związaną z tym, że nie można wszystkim pomóc, ale myślę, że trzeba o tym wiedzieć i próbować, bo są takie firmy, które nie mają przez 6 miesięcy zleceń, a mają swoje kredyty, mają swoje historie. Tak że myślę, że pytania pani poseł i pana posła Napieralskiego są absolutnie zasadne, po prostu żeby zwrócić uwagę na te firmy.

Zapraszam, panie pośle. Panie Ministrze! Pani poseł Wielichowska powiedziała, że rozumie, że jest pandemia, że tak naprawdę jest kryzys, ale zadała bardzo konkretne pytania. Proszę sobie wyobrazić, że koncert to nie tylko gwiazda, która jest na estradzie, o tym mówił również pan marszałek. Ktoś musi tę scenę zbudować, ktoś musi ją oświetlić, nagłośnić.

To jest blisko 300 tys. ludzi, którzy nie mają dzisiaj żadnych środków do życia, powtarzam: żadnych środków do życia. Rząd się nad nimi nie pochylił. Rozumiemy, że nie może być koncertów, rozumiemy, że nie może być różnych wydarzeń, ale chcemy, aby ta branża (Dzwonek), żeby ci ludzie, którzy mają rodziny i kredyty, otrzymali pomoc. Bo to nie są tylko te koncerty, które widzimy na Stadionie Narodowym, czy wielkie gwiazdy, które przyjeżdżają do nas spoza granic naszego kraju.

Oni do końca roku nie będą pracować, nie ma na to żadnych szans. Mówię: być może, bo nie wiemy, co się wydarzy. Tak wielkich przedsięwzięć nie robi się z dnia na dzień. Trzeba mieć wszystkie pozwolenia, trzeba być przygotowanym, ubezpieczonym. Panie ministrze, zapraszam. Panie Marszałku! Panie Pośle! Ja nie podważam sensowności czy zasadności tego pytania, tak samo jak nie podważam tego, że ta branża znalazła się w bardzo trudnej sytuacji.

Tylko tak jak mówię, są to obiektywne okoliczności. Nie mogę jednak zgodzić się ze stwierdzeniem, że żadnej pomocy tym ludziom nie udzielono, ponieważ tak jak mówię, oni mieli prawa do świadczenia postojowego, ciągle je mają, zostali zwolnieni ze składek ZUS.

Wręcz przeciwnie, ogromna pomoc została udzielona.

Widzę dane o programie „Kultura w sieci” z budżetem 80 mln zł, widzę gwarancje kredytowe dla sektora kreatywnego oferowane przez BGK na kwotę 500 mln zł.

Ja jako przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki też bym wolał. W ramach swoich możliwości państwo stara się wesprzeć przedsiębiorców, w tym również przedsiębiorców z tej branży.

Spotykamy się, podawałem konkretne daty spotkań pani premier. Kolejne spotkania są w planach, więc naprawdę jesteśmy w dialogu z tą branżą. To życzymy skuteczności w tym dialogu. Proszę państwa, pani poseł Barbara Bartuś z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość zada pytanie w sprawie zaawansowania prac na rzecz rozbudowy drogi krajowej nr 28 na odcinku od Nowego Sącza do Jasła, ze szczególnym uwzględnieniem planów rozbudowy ronda turbinowego w Gorlicach oraz konieczności budowy obwodnic Gorlic i Grybowa. Na to pytanie odpowie pan minister Rafał Weber, którego już raz witaliśmy. Pani poseł, bardzo proszę. Panie Ministrze! Tak jak pan marszałek powiedział, już raz witaliśmy pana ministra przy okazji odpowiedzi na poprzednie pytanie.

Inwestycje drogowe to jest też okazja do tego, aby pobudzić polską gospodarkę. Ale to jest tak, że jeżeli mówi się, że czegoś jest więcej, coś jest lepiej, to zawsze chciałoby się jeszcze więcej i jeszcze lepiej.

I właśnie o te Gorlice chciałam pana ministra w kilku słowach zapytać. Po pierwsze chciałabym zapytać o przetarg, który się już odbył, na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi krajowej nr 28 na odcinku w Gorlicach wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych i sprawowaniem nadzoru autorskiego, i dalszy możliwy termin kolejnych etapów tego zadania, czyli to przysłowiowe rondo turbinowe na Zawodziu w Gorlicach. Ale chciałabym też zapytać w kontekście odpowiedzi, którą otrzymałam w lutym, na moją interpelację w sprawie inwestycji, rozbudowy drogi krajowej nr 28 na odcinku Nowy Sącz - Ropa i rozbudowy drogi krajowej na odcinku Ropa - granice województwa małopolskiego. Pragnę zapytać właśnie o postęp tych prac w tych zadaniach, ale też o uszczegółowienie (Dzwonek) zakresu planowanych prac. Czy planowane są pasy zwalniające na podjazdach pod wzniesienia? I czy Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad w Krakowie korzysta z planów opracowywanych przez lokalne samorządy, m.in. planu budowy chodnika w Ropie i budowy ronda w Ropie? Dziękuję. Szanowni Państwo! W poprzednim wystąpieniu głównie uwagę skupiłem na inwestycjach nowych, na budowie nowych odcinków dróg szybkiego ruchu. Natomiast przy tym pytaniu pani poseł Barbary Bartuś jest dobra okazja do tego, aby powiedzieć o naszych zadaniach, które są realizowane na sieci już istniejącej, bo to też lwia część inwestycji, która jest prowadzona przez Ministerstwo Infrastruktury, a dokładniej rzecz ujmując, przez 16 oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jeżeli chodzi o drogę krajową nr 28 na odcinku małopolskim, to tak jak pani poseł wspomniała, 6 maja został ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji dla rozbudowy tej drogi na odcinku w Gorlicach.

W sierpniu tego roku, czyli w przeciągu najbliższych kilkunastu dni, dojdzie do zawarcia umowy z wykonawcą i dalsze etapy zadania, takie jak uzyskanie pozwoleń i przeprowadzenie przetargu na roboty, zostały zaplanowane tak, aby mogły się odbyć w kolejnych latach w tej perspektywie 4-, 5-letniej. Tak że jeszcze w sierpniu tego roku dojdzie do podpisania umowy, w ramach której zostanie przygotowane studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe dla odcinka drogi nr 28 w Gorlicach. Szacujemy, że wartość tego zadania będzie wynosiła 73 mln zł. Tyle jest zaplanowane w programie inwestycyjnym na to zadanie. W przypadku rozbudowy drogi krajowej na odcinku Nowy Sącz - Ropa i Ropa - granica województwa małopolskiego minister infrastruktury na przełomie poprzedniego i bieżącego roku uzgodnił programy inwestycji, a więc te zadania też zostały skierowane do realizacji. Aktualnie są one na etapie przygotowania do ogłoszenia przetargów na wykonanie dokumentacji. Tak że będą one postępowały sukcesywnie jeszcze latem tego roku. Co do zakresu rozbudów, to mają one charakter kompleksowy. Oznacza to, że na łącznie prawie 50 km drogi krajowej nr 28 od Nowego Sącza przez Grybów, Ropę, Szymbark, Gorlice aż do granicy województwa z Podkarpaciem poza podniesieniem nośności nawierzchni do 11,5 t i przystosowaniem do obowiązujących parametrów technicznych planujemy wykonać także przebudowę skrzyżowań, przebudowę mostów, przebudowę przepustów drogowych, budowę i przebudowę chodników i ścieżek pieszo-rowerowych, budowę zatok autobusowych, budowę pasów wyprzedzania, przebudowę zjazdów, wykonanie kanałów technologicznych i stabilizację osuwisk. W szczególności planowana jest budowa niezbędnych pasów wyprzedzania, przebudowa skrzyżowania drogi krajowej z drogami wojewódzkimi w Gorlicach na rondo turbinowe dwupasowe i wykonanie chodnika w Ropie. Optymalny zakres inwestycji jest opracowywany indywidualnie do potrzeb danego odcinka drogi i zgodnie z wynikami analiz stanu i bezpieczeństwa infrastruktury. Takie elementy jak pasy zwalniające na przejazdach pod wzniesienia, o które pani poseł pytała, będzie można wdrożyć na etapie sporządzenia dokumentacji. W zakresie Gorlic i Grybowa po przeanalizowaniu m.in. natężenia ruchu, wypadkowości, powiązania z drogami innych kategorii, ale także na potrzeby sieci dróg krajowych, zdecydowano, że optymalnym rozwiązaniem na najbliższe lata będzie kompleksowa rozbudowa istniejących odcinków bez zmiany przebiegu. Tak że, szanowni państwo, szanowna pani poseł, te inwestycje będą realizowane w przeciągu najbliższych lat. Program na rozbudowę drogi krajowej nr 28 w Gorlicach, tak jak powiedziałem, został oszacowany na 73 mln zł, a program inwestycyjny polegający na przebudowie tej drogi na odcinku Nowy Sącz - Ropa to blisko 200 mln zł, dokładnie 195 mln zł, i program inwestycyjny od Ropy do granicy województwa - 128 mln zł. Tak że to są te wymierne środki finansowe, które będą realizowane, można powiedzieć, że są już realizowane, po to, aby poprawić bezpieczeństwo w ruchu drogowym na drodze krajowej nr 28 we wschodniej części województwa małopolskiego. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o pytanie dodatkowe. Dziękuję. Panie Ministrze! I chciałabym zapytać znowu w kontekście tego, co mówiłam, że jeżeli coś się udaje, to dlaczego nie więcej. A więc bardzo dziękuję za to, że Limanowa czy Piwniczna znajdują się w programie budowy 100 obwodnic, ale moje pytanie: Czy w tym programie znajdą się Gorlice, mimo że tutaj przebudowujemy? Czy ta przebudowa może nie powinna być w mniejszym zakresie, a Gorlice potrzebują dużej obwodnicy? To nie jest związane z tym pytaniem, ale z moim terenem, dokładnie z Ropą, o której tutaj już była kilka razy mowa. Tam była taka przykra sytuacja (Dzwonek), że powiat zwrócił się o pieniądze, otrzymał te pieniądze, ale nie podpisał umowy. Bo to jest bardzo ważna droga i już została rozpoczęta przebudowa. Zostawiam apel, prośbę, żeby przywrócić tę drogę z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych na ten rok, bo starostwo jest gotowe na ogłoszenie przetargu już w tym momencie. Dziękuję. Proszę bardzo. Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Mamy podpisanych już ponad 70 programów inwestycyjnych, a podpisanie programu inwestycyjnego jest ni mniej, ni więcej jak tylko taką rzeczywistą decyzją o wykonaniu danego zadania, o realnym rozpoczęciu danej inwestycji. Tak że ze 100 obwodnic, które będziemy w ramach tego programu realizowali, ponad 70 programów już mamy uzgodnionych i podpisanych. Budowa obwodnicy Gorlic znajduje się w programie w załączniku nr 2. Lista rezerwowa będzie realizowana, kiedy pojawią się oszczędności poprzetargowe w ramach tych projektów, które są na liście podstawowej. Jeżeli ten trend utrzyma się przez najbliższe lata, to, jestem przekonany, wiele zadań z tej listy rezerwowej będzie realizowanych i spełnimy te oczekiwania, bardzo duże oczekiwania społeczne zarówno w Małopolsce, jak i na Mazowszu, w województwach: śląskim, świętokrzyskim, podkarpackim, we wszystkich regionach. Natomiast wracając do drogi nr 28, w ramach programu 100 obwodnic na liście podstawowej znajdują się inne obwodnice: Limanowej, Makowa Podhalańskiego, Wadowic oraz, już na Podkarpaciu, Miejsca Piastowego. Tak że widzimy ten ciąg drogowy na linii wschód - zachód na południu naszego kraju jako strategiczny i robimy wszystko, aby go udrażniać i likwidować wąskie gardła. Pytanie o Fundusz Dróg Samorządowych. To zagadnienie, które pani poseł poruszyła, jest analizowane od strony prawnej.

Zobaczymy, do czego nas obliguje ustawa o Funduszu Dróg Samorządowych i w jaki sposób ten problem można rozwiązać.

Te środki, tak jak pani poseł powiedziała, zostały skierowane na inne zadania z listy rezerwowej Funduszu Dróg Samorządowych. Zobaczymy, jak ta lista, i powiatowa, i gminna, będzie konsumowana, ile tych oszczędności będzie się pojawiało w ramach innych przetargów. Mamy relacje ze wszystkich województw, że te oszczędności naprawdę są [[Dzwonek]] - czasami to są oszczędności rzędu nawet 30% - tak że kolejne zadania z listy rezerwowej wchodzą i są dofinansowywane. Będziemy tutaj działać na gruncie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych.

Ale pan minister za chwilę będzie mógł jeszcze kilka słów powiedzieć na tematu budowy drogi Via Carpatia, gdyż w tej sprawie posłowie Jerzy Paul, Adam Śnieżek oraz Piotr Uruski, przedstawiciele Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, zadadzą panu ministrowi pytanie.

Chciałbym zadać pytania w sprawie, która interesuje nie tylko moich wyborców, ale też znaczną część mieszkańców Unii Europejskiej. Chodzi o drogę Via Carpatia, która ma przebiegać przez Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię i Grecję, stanowiąc szlak transportowy prowadzący wzdłuż granicy wschodniej Wspólnoty Europejskiej.

Jak sytuacja zagrożenia epidemiologicznego związana z wirusem COVID-19 wpłynęła na przebieg inwestycji i czy były odcinki, na których prace zostały wstrzymane? Na ile odcinków są podpisane umowy o realizację, a na ile - rozpisane przetargi? Czy przewidywany termin zakończenia tej niezwykle ważnej inwestycji nie jest zagrożony? Dziękuję za uwagę. Dziękuję serdecznie. Zapraszamy pana ministra. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pan marszałek kilkanaście minut temu stwierdził, że aż ma ochotę wyjechać i ruszyć w teren, ruszyć w Polskę.

Teraz sprawdzam na nawigacji. Podróż z Warszawy do Ustrzyk to w tej chwili 6 godzin 20 minut, natomiast po wybudowaniu Via Carpatii, szczególnie tych odcinków między Lublinem a granicą ze Słowacją, sądzę, że ta podróż skróci się, przy swobodnej jeździe zgodnie z prawem, do 4 godzin. Trzeba podkreślić, że jest ona realizowana właśnie dzięki konsekwentnej polityce Prawa i Sprawiedliwości, polityce realizowanej od wielu, wielu lat. Inicjatorem idei budowy Via Carpatii jako szlaku o międzynarodowym znaczeniu był śp. prezydent Polski pan prof. Lech Kaczyński. Przypominam rok 2006 i spotkanie w Łańcucie z przedstawicielami Litwy, Słowacji i Węgier. Wtedy cztery państwa wyraziły zainteresowanie budową tego szlaku. W tej chwili - po zabiegach, tak jak powiedziałem, w głównej mierze polityków Prawa i Sprawiedliwości, także tych związanych z województwem podkarpackim, pana europosła Tomasza Poręby, pana marszałka Marka Kuchcińskiego, ale też po przejęciu władzy w roku 2015, po zapewnieniu finansowania budowy tej drogi, bo to, przypominam, decyzja rządu jeszcze pani premier Beaty Szydło z roku 2017 zapewniła finansowanie Via Carpatii - tą drogą interesuje się już 12 państw, od Litwy poprzez Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię, Grecję, ale także kraje takie jak Chorwacja, Serbia, Czarnogóra, czyli kraje bałkańskie. I cieszę się bardzo, naprawdę, panie marszałku, że nam przychodzi realizować ten projekt. Na szczegółowe pytanie pana posła odpowiem w formie pisemnej. Mogę tak bardzo ogólnie powiedzieć, że odcinki S19 na terenie województwa podkarpackiego na północ od Rzeszowa to jest sześć odcinków realizacyjnych. Wszystkie są już w fazie prac ziemnych. Rok 2021 - zgodnie z harmonogramem oddanie czterech z nich.

W trakcie przygotowywania procesów przetargowych są kolejne odcinki. Tak że te przetargi będą ogłaszane, umowy będą podpisywane, inwestycja będzie realizowana, a na tym terenie województwa podkarpackiego naprawdę ona wymaga dużej sprawności budowlańców. Tam będą bardzo długie tunele. Dość powiedzieć, że szacujemy, że odcinek między Rzeszowem a Barwinkiem o długości blisko 90 km będzie polskie państwo kosztował 11 mld zł. Uznajemy tę drogę za strategiczną nie tylko dla takich regionów jak Podkarpacie, Lubelszczyzna czy Podlasie, ale to jest naprawdę szlak o międzynarodowym znaczeniu i środki finansowe na tę drogę musiały zostać znalezione i zostały w roku 2017 znalezione, a przy ostatniej nowelizacji programu budowy dróg krajowych i kolejnym podniesieniu limitu, widząc sytuację poprzetargową, również na ten odcinek południowy, ale też na odcinek między Lublinem a Białymstokiem przeznaczyliśmy kolejne miliony złotych, w zasadzie miliardy złotych, aby na tę inwestycję środków finansowych nie brakowało. Jeszcze raz dziękuję wszystkim tym, którzy dbali o to, aby Via Carpatia była na agendzie międzynarodowej. Dziękuję tym, którzy później już, mając możliwości decyzyjne, podejmowali decyzje o zabezpieczeniu finansowym, bo dzięki temu teraz możemy tę drogę (Dzwonek) realizować. Dziękuję, panie ministrze. Panie pośle, czyli jest dobrze. Proszę bardzo. Jeszcze jedno pytanie.

Myślę, że tak, ale posłuchamy za chwilę. Wysoka Izbo! Tak jak powiedziałem, kilka dni temu doszło do podpisania umowy na jeden z pięciu odcinków realizacyjnych. Są przygotowywane teraz postępowania przetargowe na cztery kolejne odcinki realizacyjne. Tak że mamy ponad 5 lat, 6 lat na wybudowanie Via Carpatii między Rzeszowem a granicą ze Słowacją. Tak jak powiedziałem wcześniej, to są bardzo trudne odcinki od strony techniczno-inżynieryjnej. Tunele, które będą prowadziły pod górami, pod terenami województwa podkarpackiego, wymagają naprawdę bardzo dużej precyzji i bardzo dużego doświadczenia, ale jesteśmy przekonani, że branża budowlana z tymi zagadnieniami sobie poradzi. Politycy swoje zrobili. Politycy znaleźli finansowanie, politycy zagwarantowali środki finansowe, natomiast teraz wszystko w rękach budowlańców. Jesteśmy przekonani, że budowlańcy z tym zagadnieniem sobie poradzą. A mówiłem wcześniej o tym, że politycy Prawa i Sprawiedliwości nie tylko interesują się Via Carpatią, ale też dokonali wymiernych działań, aby tę drogę zrealizować. Przykład tej dyskusji jest też znaczący.

Są ważniejsze rzeczy do realizacji. To świadczy o tym w sposób bardzo dobitny. Mamy nadzieję, że wszystkie harmonogramy, wszystkie terminy, które są teraz założone, zostaną dotrzymane. Do widzenia. Posłowie Marek Polak oraz Krzysztof Tchórzewski z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość chcieli zadać pytanie w sprawie efektów wprowadzenia tarczy antykryzysowej dla małych i dużych przedsiębiorstw. Na to pytanie będzie odpowiadał podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju pan minister Marek Niedużak.

Witam serdecznie. Dziękuję bardzo. Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Z informacji przekazanych przez Ministerstwo Rozwoju wynika, że pierwsze dni pandemii koronawirusa wywołały falę zawieszania i zamykania przedsiębiorstw oraz pojawił się zamiar znacznej redukcji zatrudnienia. Sytuacja ta zaczęła się dopiero stabilizować wraz z wprowadzeniem poszczególnych etapów tarczy antykryzysowej oferującej przedsiębiorcom różnorodne wsparcie ze strony państwa. Z danych Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wynika, że w marcu br. swoją działalność zawiesiło blisko 49 tys. firm, a w kwietniu niemal 24 tys., czyli aż o 50% mniej. I chciałbym zapytać, jaki wpływ mają mechanizmy wprowadzane w ramach tarczy antykryzysowej na powstrzymanie niepokojącego zjawiska zawieszania i likwidowania przedsiębiorstw i czy dzięki przekazanemu wsparciu udało się ograniczyć redukcję zatrudnienia w polskich zakładach pracy. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Proszę, panie ministrze.

Wysoka Izbo! Panie Pośle! Chciałbym zacząć od informacji o tym, że liczba wniosków o zawieszenie i zakończenie działalności gospodarczej według stanu na dzień 13 lipca to było 8,3 tys. i to była liczba o 12% niższa w stosunku do tego samego okresu w poprzednim miesiącu i o 53% niższa niż rok temu. Co więcej, kiedy popatrzymy na liczbę podmiotów, liczbę przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG, w centralnej ewidencji, to dziś mamy ich zarejestrowanych więcej niż przed pandemią, czyli obserwujemy na poziomie centralnej ewidencji, z jednej strony, zmniejszającą się liczbę wniosków o zawieszenie i zakończenie działalności gospodarczej, ona spada, spada liczba tych wniosków, a z drugiej strony, mamy więcej przedsiębiorców aktywnych w CEIDG, więcej niż przed pandemią. To jest oczywiście bardzo dobry sygnał. To pokazuje, że stopniowo polska gospodarka odmraża się, wraca do aktywności, wraca do życia. I to pokazuje, że zasadniczo ten kierunek odmrażania gospodarki, przynajmniej z tej perspektywy, z perspektywy gospodarczej, jest jak najbardziej słuszny, uzasadniony. Należy pamiętać, że tutaj bardzo istotna jest kwestia spraw epidemiologicznych, sanitarnych, które są decydujące, powinny być decydujące.

I teraz, czy te pozytywne dane w jakiś sposób są powiązane z pomocą udzielaną przez państwo? Powiem tak, tak się złożyło szczęśliwie, choć mam przygotowany też materiał, że dzisiaj nawet natknąłem się w prasie na materiał, który, wydaje mi się, idealnie wpisuje się w to pytanie i dlatego pozwolę sobie z niego skorzystać.

I tutaj przedstawiciele tej branży wyraźnie mówią o tym, że mamy pozytywne zjawisko w postaci braku zatorów płatniczych. Widzimy pewne opóźnienia w płatnościach, ale skala ich była niewielka. I widzimy u przedsiębiorców zapasy gotówki. Tu wręcz cytuję artykuł i wręcz cytuję przedstawicieli tej branży: zapasy gotówki pochodzące z transferu z PFR przekazywane w ramach tarczy finansowej.

I tutaj zwróćmy uwagę chociażby na aktywność BGK, na gwarancje de minimis, ale również na takie elementy regulacyjne, bo chociażby w pierwszej ustawie, którą potocznie nazywamy tarczą, również były przepisy, które, wprost powiedzmy, zachęcały banki do nieodcinania przedsiębiorców od kredytu obrotowego.

A właśnie przecież sytuacja płynnościowa to jest właśnie to, co się bezpośrednio przekłada na to, czy przedsiębiorca, nie wiem, w skrajnym wypadku składa wniosek o upadłość albo tak jak tutaj w pytaniu padło, chce zawiesić działalność gospodarczą czy też z niej w ogóle zrezygnować, wnosząc o wykreślenie z ewidencji.

Dziękuję. Pytanie dodatkowe, pan poseł Marek Polak. Dziękuję bardzo. Panie Ministrze! Z chwilą pojawienia się pandemii i problemów z nią związanych aż 28% firm wprost deklarowało, że aby przetrwać, musi bezwzględnie zredukować zatrudnienie. Proszę powiedzieć, czy wprowadzone rozwiązania w ramach tarczy antykryzysowej zmniejszyły ten odsetek i czy dużo jest przedsiębiorstw, które pomimo oferowanej pomocy ze strony państwa nie poradzą sobie ze skutkami tego kryzysu. Dziękuję bardzo.

Wysoka Izbo!

Natomiast nic dzisiaj nie wskazuje na to, że ono się zwiększy w sposób dramatyczny. Miliony polskich pracowników, czy mówiąc troszkę mniej, że tak powiem, osobowo, miliony miejsc pracy są objęte pomocą oferowaną czy to w ramach tzw. przestoju ekonomicznego, czy w ramach pomocy, do której przedsiębiorcy czy pracodawcy mają dostęp ze względu na to, że mają obniżone obroty, czy to w ramach tarczy finansowej, środków, które przedsiębiorcy mogli pozyskać za pośrednictwem PFR-u, sieci banków komercyjnych.

Bezrobocie w Polsce mamy obecnie na poziomie 6,1%.

Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie panu ministrowi. Pytanie to kończy rozpatrywanie tego punktu porządku dziennego, ale zanim przejdziemy do punktu 18., musimy ogłosić przerwę, gdyż nie ma wnioskodawcy.

Jest wnioskodawca. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 18. porządku dziennego: Informacja bieżąca. Przypominam, że na obecnym posiedzeniu Sejmu zostanie rozpatrzona informacja w sprawie zaangażowania instytucji państwa w proces wyborczy w czasie wyborów prezydenta RP, w tym organizacji wyborów przez MSZ, wykorzystania alertu RCB rozsyłanego przed drugą turą wyborów oraz zaangażowania mediów publicznych, o której przedstawienie wnosił Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni. Przypominam również, że przedstawienie uzasadnienia wniosku przez posła przedstawiciela wnioskodawców nie może trwać dłużej niż 5 minut, a udzielenie odpowiedzi przez przedstawiciela Rady Ministrów - dłużej niż 5 minut. Wystąpienia posłów w dyskusji nie mogą trwać dłużej niż 2 minuty. Na zakończenie dyskusji głos zabierają kolejno przedstawiciele wnioskodawców oraz przedstawiciel Rady Ministrów. Wystąpienie przedstawiciela wnioskodawców nie może trwać dłużej niż 5 minut, a wystąpienie przedstawiciela Rady Ministrów - dłużej niż 5 minut. Marszałek Sejmu może wyrazić zgodę na wydłużenie wystąpienia przedstawiciela Rady Ministrów. Czas przeznaczony na rozpatrzenie punktu: Informacja bieżąca nie może być dłuższy niż 90 minut. Proszę bardzo, panie pośle. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ten punkt, rozpatrywany przy nieco pustej ławie Rady Ministrów, jest bardzo ważny, jeśli patrzymy na to, w jaki sposób te wybory były zorganizowane, jak nieuczciwie. Szanowni państwo, wykorzystaliście aparat państwowy do tego, by wybory nie były równe i nie były powszechne. Dopuściliście się wielu nadużyć, które w naszej ocenie mogły wpłynąć na wynik wyborczy, i pokrótce udowodnimy, jakie to były kwestie. Od samego początku - po pierwsze, przyjęliście zmiany w prawie wyborczym w sposób niezgodny z polską konstytucją. Po drugie, przeznaczyliście dla kandydatów nierówne limity finansowe, co w sposób oczywisty rzutowało na sposób prowadzenia kampanii. Ale stały się rzeczy dużo bardziej poważne. Wykluczyliście swoją nieudolnością i niewłaściwym działaniem aparatu państwowego dziesiątki tysięcy osób z procesu wyborczego, w szczególności mam na myśli osoby, które nie mogły zagłosować za granicą. W dodatku oszukiwaliście opinię publiczną, chociażby w stosunku do osób, które mieszkają w Irlandii. Mówiliście, że tam nie można osobiście odbierać pakietów wyborczych. Tymczasem na skutek opóźnień setki, tysiące osób nie oddały głosu w tych wyborach. Dlaczego te wybory były nieuczciwe? Cały aparat państwowy w sposób niezgodny z prawem został zaangażowany do promocji jednego kandydata - obecnie urzędującego prezydenta Andrzeja Dudy. Premier Mateusz Morawiecki, zamiast zajmować się zarządzaniem krajem, zamiast zajmować się organizacją pracy Rady Ministrów, zajmował się wiecami Andrzeja Dudy. W dodatku rozdawał czeki bez pokrycia, bo przypomnę, że ten cyrk, który urządziliście w całym kraju, nie miał podstaw prawnych. Rozdawaliście pieniądze, których nie ma ani w budżecie, ani nie było w ogóle podstaw prawnych, bo ustawa nie była przyjęta. Strony internetowe urzędów wojewódzkich były pełne informacji na temat kandydata na prezydenta, które nie były związane z wykonywaniem przez niego mandatu prezydenta Rzeczypospolitej. Wreszcie rzecz absolutnie niedopuszczalna - bezprawnie użyliście systemu RCB, który jest po to, by ostrzegać ludzi przed niebezpieczeństwami, użyliście go do propagandy wyborczej, niestety, w sposób bezprawny. I kolejna rzecz niedopuszczalna - chyba każdy z kandydatów partii opozycyjnych, każdy z kandydatów innych komitetów doznał niesamowitego hejtu, manipulacji i kłamstw ze strony mediów państwowych, na które najpierw przeznaczyliście 2 mld zł. Osobiście za to odpowiada ten rząd, osobiście za to odpowiada większość parlamentarna, ale również prezydent Rzeczypospolitej. Urządziliście rzecz, która wcześniej w wolnej Polsce była rzeczą nie do obrony, a mianowicie cała propaganda państwowa została użyta do tego, by z jednej strony bez wskazania źródła finansowania propagować jednego kandydata, pomagać mu, a z drugiej strony stworzyliście machinę hejtu i nienawiści wymierzoną w innych kandydatów. Stworzyliście mechanizm, który ma wam zapewnić kolejne wygrywanie wyborów. I dzisiaj ta informacja ma właśnie pokazać opinii publicznej, że jesteście ludźmi skrajnie nieuczciwymi. Nie potraficie zmieścić się w zasadach demokracji parlamentarnej i standardach demokratycznych, bo wiecie, że w normalnych warunkach byście przegrywali. I to nie jest tak, że my wam zarzucamy fałszerstwa wyborcze. W Rosji, w krajach niedemokratycznych też fałszerstw nie ma, tam po prostu się eliminuje konkurentów. Wy jeszcze nie jesteście na etapie wsadzania do więzień, tak jak w tzw. demokracjach wschodnich, kandydatów, żeby nie mogli startować, ale aparat państwowy zaangażowaliście do tego, by zdyskredytować kandydatów. Kiedy mówimy o tych wszystkich nieprawidłowościach, raz jeszcze chcemy podkreślić: Wybory nie były równe i nie były powszechne, wybory były nieuczciwe. I my upominamy się o elementarną przyzwoitość, o to, by pokazać opinii publicznej, w jaki sposób cały aparat państwowy nielegalnie został zaangażowany po stronie jednego kandydata - urzędującego prezydenta. Kłamaliście, kłamiecie i będziecie kłamać. I niestety to jest dewiza obecnej władzy. Dziękuję serdecznie. Będę prosił w kolejności o udzielenie odpowiedzi panów: sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych pana ministra Piotra Wawrzyka, następnie sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji pana Pawła Szefernakera i następnie sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego pana Pawła Lewandowskiego. Przypominam uprzejmie i grzecznie trzem panom, że łącznie macie 5 minut. Zapraszam pana Piotra Wawrzyka.

Gratuluję wystąpienia panu przewodniczącemu. Widać, że mówił znawca tematu.

Proszę popatrzeć, ile osób wtedy brało udział w wyborach, a ile teraz brało udział w wyborach.

178 to były te niedoręczone. To gdzie te setki tysięcy, które zostały pozbawione prawa udziału w wyborach? A dlaczego tak się stało? To była ta sytuacja, o której pan powiedział.

I to, można powiedzieć, że jest droga uprawniona, tylko że zwrócił się do ministerstwa do spraw dzieci, które ma niewiele wspólnego ze zgodą wydawaną państwom trzecim, jak Polska, na organizację w tym kraju wyborów. Myśmy się trzy razy zwracali w Irlandii do ministerstwa spraw zagranicznych, które w tym zakresie jest partnerem, i trzy razy dostawaliśmy noty stwierdzające, że nie jest możliwy osobisty kontakt ze względu na dużą liczbę osób zarejestrowanych, zwracam uwagę, 30 tys.

To będzie właśnie ta sytuacja z tzw. zabójczymi kopertami, o których mówiliście państwo, nie chcąc dopuścić do wyborów 10 maja. To wtedy właśnie byłyby te zabójcze koperty, gdyby zrobić to, czego chcieliście, w Irlandii, zresztą w innych krajach również.

Wiem, że to pana może śmieszy, panie pośle, ale tak niestety było. Ja to rozumiem. Dla mnie to jest powód do dumy, że mimo to udało się tak sprawnie te wybory przeprowadzić. Że 86% tych, którzy chcieli brać udział w wyborach, w tych wyborach wzięło udział, że 86% wyniosła frekwencja.

Dziękuję serdecznie.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Spróbuję się pilnie odnieść do jednej kwestii, do której zostałem upoważniony przez Radę Ministrów, chodzi o alert RCB. W rozporządzeniu ministra zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanych ze zwalczaniem epidemii COVID dla członków obwodowych komisji wyborczych wprowadzono przepisy istotne z punktu widzenia zagrożenia epidemicznego. Dzięki tej nowelizacji na kilka dni przed drugą turą wyborów pierwszeństwo w obsłudze podczas wyborów uzyskały osoby z grup szczególnie wrażliwych (Dzwonek), m.in. seniorzy, kobiety w ciąży czy osoby z niepełnosprawnościami. Przepisy te weszły w życie kilka dni przed drugą turą wyborów. 2 dni przed wyborami Państwowa Komisja Wyborcza zaapelowała w komunikacie do organów władzy i administracji publicznej o jak najszersze rozpowszechnienie wśród wyborców informacji o zmianie zasad obsługi przez obwodowe komisje wyborcze. Alert RCB umożliwia szybkie dotarcie do szerokiego grona odbiorców. W związku z tym apelem PKW wykorzystano to do rozpowszechnienia informacji o zmianie prawa. Chciałbym w tej chwili zaznaczyć, że alert RCB kilkukrotnie był używany w celu powiadomienia obywateli o nowych przepisach związanych z zagrożeniem koronawirusem. SMS-y dotyczące m.in. wprowadzenia obowiązku zakrywania nosa, ust czy znoszenia kolejnych obostrzeń wynikających ze zmiany rozporządzeń Rady Ministrów wysyłano w marcu i kwietniu tego roku kilkukrotnie.

Kompletnie chciałbym się z tym nie zgodzić, panie przewodniczący. W alercie była informacja o zmianie prawa związanej z sytuacją epidemiczną. To po pierwsze. Nie było tam nic, co miałoby znamiona tego, o czym pan mówi. Chciałbym skończyć, cytując byłego szefa PKW pana Wojciecha Hermelińskiego, który pytany przez Onet o decyzję RCB, odpowiedział: Nie kwestionowałbym tego rozporządzenia z prawnego punktu widzenia.

Dziękuję serdecznie.

Mamy prezydenta. Opozycja przegrała te wybory, ale kurz kampanii jeszcze nie opadł, no i nie może się pogodzić się z przegraną. Podmienionym kandydatem Koalicji Obywatelskiej, a tak chciałoby się powiedzieć, polskiej partii uczciwości, został prezydent Warszawy ledwie 1,5 roku wcześniej wybrany na tę funkcję. Zamiast zajmować się sprawami stolicy i jej mieszkańców, zostawił wszystko na pastwę losu i pojechał w Polskę robić kampanię wyborczą. A co tymczasem w Warszawie? Wspomnę tylko o wypadkach autobusów miejskich. 25 czerwca - tragiczny wypadek na moście Grota-Roweckiego. 22 osoby ranne, jedna nie żyje. 7 lipca - kolejny wypadek. Autobus zjeżdża z drogi i taranuje auta na Bielanach. Mam w związku z tym pytanie: Pod czyim nadzorem znajduje się transport miejski w Warszawie? Kto zdecydował, że usługi autobusowe wykonuje niemiecka spółka Arriva? Czy półetatowy prezydent ocknie się w końcu i zajmie się tym, co do niego należy? Dziękuję serdecznie. Proszę pana, lista osób oczekujących na zabranie głosu została ustalona. Wpisaliście się państwo w takiej kolejności. Panie Marszałku!

Kłamiecie rano, kłamiecie w południe i potraficie kłamać wieczorem. Pan prezydent obiecał, że Kurskiego wyrzuci. Kurski ma się dobrze. Notabene wczoraj przychodzi do pana marszałka Terleckiego z prywatną wizytą, chyba - nie wiem - omawiać sukcesy tej kampanii wyborczej. A wy tutaj wyjeżdżacie z autobusami w Warszawie. To pokazuje stan waszego umysłu. Nie potraficie powiedzieć: przepraszam, wygraliśmy nieuczciwie, dlatego że raz zdobytej władzy nie chcemy oddać. Ale Polakom należy się jasne wytłumaczenie. Stworzyliście system, który ma gwarantować tę medialną otoczkę nad waszymi kłamstwami. Nie potrafiliście przeprowadzić uczciwej, rzetelnej dyskusji o Polsce. Zastąpiliście to telewizją Kurskiego i 2 mld zł, które zabraliście obywatelom. Zabraliście pieniądze, które mogły iść na służbę zdrowia, a poszły na propagandę.

Bo tam mają was po prostu dosyć i przyszli głosować przeciwko wam. A wy zrobiliście wszystko, żeby te osoby nie mogły zagłosować. Pani posłanka Katarzyna Kretkowska, klub parlamentarny Lewica. Wysoka Izbo! Klub parlamentarny Lewicy niezależnie od tego, kto wygrał wybory, kto je przegrał, jest w dyskusji nad samym przebiegiem wyborów przede wszystkim zainteresowany tym, czy każda Polka i każdy Polak byli potraktowani podmiotowo i mieli szansę oddać głos. Pierwsza kwestia dotyczy głosowania w DPS-ach. Pojawiają się informacje medialne pokazujące, iż w niektórych DPS-ach 100% osób oddało głos na jednego kandydata. To nie jest tak, że to było powszechne i we wszystkich DPS-ach, niemniej w wielu DPS-ach tak było.

Druga kwestia dotyczy głosowania za granicą. Na podstawie lektury tego, o czym pisały same konsulaty polskie za granicą, nie ma podstaw, ażeby mieć pretensje do pracy tych konsulatów, o czym zresztą mówił pan minister, bo wydaje się, po prześledzeniu tego, co same konsulaty publikowały na swoich stronach, że dołożyły one wszelkich starań, ażeby w drugiej turze otrzymane pakiety, wzory kart do głosowania wydrukować i wysłać w możliwie najszybszym czasie - 24 godzin.

W związku z tym mam pytanie: Ile jest zażaleń dotyczących niemożności oddania głosu i co rząd zamierza zrobić na przyszłość? Ja już kończę. nie zadziałało. Wydaje się, że po prostu powinno być umożliwione głosowanie elektroniczne w tej sytuacji, że ten system, który obowiązywał między pierwszą a drugą turą, jest zbyt archaiczny jak na dzisiejszy czas. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Spróbujemy się połączyć. Dobrze, łączenie nie zadziałało. W związku z tym poprosimy pana posła Sławomira Nitrasa z Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska. Ja się nawet cieszę, że to akurat pan Szefernaker w imieniu rządu tutaj występuje, bo pamiętam jego rolę w roku 2015.

Raport OBWE mówi, panie ministrze Szefernaker, że spowodowaliście zatarcie granic pomiędzy państwem a partią, co stworzyło nieuzasadnioną przewagę prezydenta ubiegającego się o reelekcję. Raport OBWE stawia nas dokładnie w tym samym szeregu co państwo Putina, bo dokładnie w tym kierunku idziecie i tak robicie wybory. Do dnia wyborczego nie można się przyczepić - każdy może przyjść i zagłosować - ale całe państwo zostało zaprzęgnięte po to, żeby wygrał pan Duda. Czy tylko urzędy wojewódzkie? O roli telewizji będziemy jeszcze dużo mówić. Poczta Polska, PKP, ulotki w pociągach - tego nigdy nie było. To jest hańba. Posunęliście się tak daleko, jak musieliście się posunąć, żeby wygrać te wybory. Jeżeli ktoś nie postawi temu tamy, to w następnych wyborach posuniecie się jeszcze krok dalej, jeżeli będzie taka potrzeba. Jeden z pana protektorów, pan Brudziński, powiedział, i ja się z nim zgadzam, że Duda wygrał wybory dzięki Kaczyńskiemu. To jest prawda. Wiecie dlaczego? Dlatego że to Kaczyński uparł się, że Jacek Kurski ma być szefem telewizji, a bez telewizji nigdy tych wyborów byście nie wygrali. Bezczelny Kurski przychodzi do Sejmu i mówi, że czas poświęcony Trzaskowskiemu był taki sam jak czas poświęcony Dudzie. To jest hańba. Kandydata, na którego głosuje 10 mln ludzi, rządowa telewizja nazywa zdrajcą, mówi, że sprzeda Polskę. Jesteście kłamcami (Dzwonek), a na czele tego aparatu postawiliście młodego, niedoświadczonego człowieka, który jedyne, co potrafi, to kłamać. Dziękuję serdecznie, panie pośle. Poprosimy panią posłankę Barbarę Dziuk, bo właśnie

Niestety moja zapowiedź nie była zgodna z prawdą. Proszę bardzo. Panie Marszałku! Wysoki Sejmie!

Rzeczywiście nigdy nie było takiego zaangażowania rządu, struktur państwa, wojewodów w kampanię wyborczą. Ale państwo poszliście dalej. Użyliście w kampanii mundurów, co jest już w ogóle niewybaczalne. Szefowie służb, Państwowej Straży Pożarnej jeździli z promesami, organizowali pokątne spotkania ze strażakami, wręczając im te promesy na samochody pożarnicze, jakby nie można było tego uczynić w sposób cywilizowany. To oczywiście kolejny krok. Działanie premiera Rzeczypospolitej Polskiej bez podstawy prawnej, tworzenie przyrzeczeń publicznoprawnych w postaci kartoników dla samorządów. Byłaby prokuratura, byłaby RIO, byłyby inne rzeczy. Ci, którzy postępują zgodnie z prawem, płacą abonament radiowo-telewizyjny, pytają: Jakim prawem jedna formacja zawładnęła telewizją publiczną i prowadziła kampanię na rzecz jednego kandydata? Odpowiedź jest taka, że to telewizje prywatne robiły, inaczej. Tylko że telewizje prywatne nie żyją z abonamentu i 2 mld zł z budżetu państwa. Żyją z reklam. Jeśli dalej tak będziecie postępować z telewizją publiczną, to nie dziwmy się, że nie będzie chętnych do płacenia abonamentu. Dziękuję serdecznie. Pan poseł Marek Polak, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Proszę bardzo, panie pośle.

Zapraszamy panią posłankę Barbarę Nowacką, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Wybory to święto.

To święto popsuliście, panie i panowie z PiS. Popsuliście je w sposób niegodny i obrzydliwy, bo te wybory nie były ani uczciwe, ani równe. To, co się udało, to wielkie poruszenie obywatelek i obywateli, to, że mimo seansów pogardy i nienawiści w TVP, mimo ulotek roznoszonych przez Pocztę Polską poszli do wyborów. Chciałam podziękować tym wszystkim, którzy nie dali się omamić i mieli odwagę pilnować tych wyborów jako mężowie i żony zaufania. Mieli odwagę patrzeć wam na ręce pomimo zastraszania. Mieli odwagę.

Nie jest wam wstyd, że przez kilka miesięcy oglądaliśmy kampanię nienawiści, wykluczającą nie tylko Rafała Trzaskowskiego, ale każdą osobę, która odważa się myśleć inaczej? Ministrowie i premierzy, ja nie mówię o politykach, ministrowie i premierzy. Premier - 200 spotkań kampanijnych, Kancelaria Prezydenta - zaangażowana w kampanię. Czy byli na urlopach? Czy wreszcie doczekamy się odpowiedzi - bo nie doczekaliśmy się odpowiedzi - kto finansował 200 agitacyjnych spotkań Mateusza Morawieckiego, kto finansował agitacyjne spotkania w OSP? Jarosław Kaczyński powiedział, że użyje wszystkich środków. I wiecie, co jest najbardziej niegodne? To, że użyliście ich dokładnie wszystkich. W domach pomocy społecznej i w zakładach, gdzie leżą osoby chore, często niepełnosprawne - 100% frekwencji i 100% na Andrzeja Dudę. To jest po prostu niegodne działanie. Jest kilkadziesiąt [[Dzwonek]] takich przypadków.

A dzisiaj strażacy w takim Orlu na Pomorzu zbierają złom, żeby kupić wóz strażacki, bo tam wasz Mateusz Morawiecki nie dojechał, bo na Pomorze się baliście. Bardzo proszę, pani poseł Barbara Bartuś, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowna Platformo Obywatelska i panie przewodniczący wnioskodawco tej informacji, boli, oj, boli ta przegrana. Ale szanowni państwo, korzystając z okazji, chciałam podziękować wszystkim tym, którzy poszli do wyborów, do wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, najważniejszych wyborów, wyborów, w których wybraliśmy głowę państwa na następne 5 lat, i oczywiście dziękuję szczególnie tym, którzy zagłosowali na Andrzeja Dudę i na kontynuację Polski+. Boli - wszystkie wozy strażackie, które były rozdawane, bo za waszych czasów to cała Polska nie miała rocznie tyle nowych samochodów strażackich co za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości.

I żadnego województwa, pani poseł, się nie baliśmy. Niezależnie od tego, w jakim województwie, jaka gmina, na kogo głosowała, jeżeli była wysoka frekwencja, to otrzymuje wóz strażacki. A jeżeli mówimy o kłamstwach i manipulacjach, szanowni państwo, i o nienawiści, to tę nienawiść widać nawet u państwa dzisiaj, kiedy szykanujecie wyborców Prawa i Sprawiedliwości i wszystkich tych, którzy głosowali na pana prezydenta Andrzeja Dudę, wymyślacie im. To z waszej strony kłamliwe oszczerstwa wprost zamieszczała prasa, ale też telewizja, jedno medium naprzeciwko drugiego. Polacy nie dali się zwieść i wiedzą, że to, że im się żyje lepiej, to dzięki współpracy rządu polskiego. na czele z panem Mateuszem Morawieckim i [[Dzwonek]] dzięki panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie, któremu też przy tej okazji w imieniu wyborców z mojego okręgu serdecznie dziękuję. Dziękujemy serdecznie. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Powracając do wystąpienia pana ministra Szefernakera, chciałbym sprostować parę informacji. Otóż wcześniejsze informacje RCB dotyczyły życia i zdrowia Polaków. Tymczasem inkryminowany SMS wysłany przez RCB dotyczył wyłącznie zmiany sposobu wejścia do lokalu, to nie było nic związanego ze zdrowiem i życiem Polaków, podczas gdy ustawa o zarządzaniu kryzysowym wyraźnie określa, że te komunikaty mogą dotyczyć wyłącznie sytuacji potencjalnych zagrożeń. To było złamanie ustawy. I kiedy wczoraj zarzuciłem to panu ministrowi Kamińskiemu, mówiąc, że kupczyliście bezpieczeństwem Polaków w trakcie wyborów prezydenckich, to pan minister powiedział, że on przecież nie ma nic wspólnego z RCB. To po prostu było wprowadzenie w błąd Wysoką Izbę, ponieważ pan minister nadzoruje, owszem, jest podporządkowane premierowi. Ale chciałbym powiedzieć o czymś innym. Chcę powiedzieć o tym, że w tych wyborach jedyną instytucję, która się cieszy powszechnym szacunkiem i sympatią, i zaufaniem Polaków, którą wyście stworzyli, czyli alert RCB, poświęciliście po to, żeby zwiększyć szanse własnego kandydata. Nie jesteście w stanie się powstrzymać w destrukcji państwa. nawet w tych sprawach, któreście sami dobrze wykonali. Jeśli dzisiaj mówimy o tych skandalicznych sprawach, to mówimy nie dlatego, że my podważamy wynik wyborów, tylko zwracamy uwagę na to, że to były wybory nieuczciwe, nierówne i niepowszechne. I robimy to dlatego, żeby nie dopuścić do dalszych waszych fałszerstw, kłamstw i manipulacji w trakcie następnych wyborów. Dziękuję serdecznie. Przeprosimy panią poseł Beatę Strzałkę, gdyż połączyliśmy się z panem posłem Markiem Polakiem. Dziękuję bardzo. Wysoka Izbo! Ja w swojej wypowiedzi chciałbym nawiązać do bezpodstawnie w mojej ocenie podnoszonego do rangi problemu faktu wykorzystania alertu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przed drugą turą wyborów. Myślę, że w czasie panującej pandemii w trosce o zminimalizowanie ryzyka zakażenia wśród dzieci, kobiet w ciąży i osób starszych nie tylko wspomniany alert, ale i wszystkie inne dostępne instrumenty i narzędzia powszechnego powiadamiania powinny być wykorzystane. Informacje o obowiązkowym zasłanianiu nosa, a także o zasadach sanitarnych obowiązujących w lokalach wyborczych powinny w każdy możliwy sposób w mojej ocenie dotrzeć do każdego wyborcy, bo mogą uratować ludzkie zdrowie, a nawet życie, co, jak wiadomo, jest wartością nadrzędną. I dziwię się, że ktoś może podnosić to do rangi problemu, co w moim przekonaniu jest czymś absolutnie niedorzecznym. Chciałbym zapytać pana ministra, czy istnieją regulacje prawne ograniczające stosowanie tego rodzaju praktyk. Zapraszam panią poseł Beatę Strzałkę z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Muszę przyznać rację pani poseł Nowackiej, bo wybory to rzeczywiście święto demokracji, ale po raz kolejny przybrały formę igrzysk, swoistego plebiscytu kandydatów. Zawsze wygrywa najlepszy. Tym razem wybory to również maraton, długi maraton, ale Andrzej Duda pokonał kontrkandydatów w sztafecie. Bo jak inaczej nazwać kampanię i zmianę kandydatki Koalicji Obywatelskiej w trakcie tej kampanii? Trudno pogodzić się z porażką. Szukacie usprawiedliwienia przegranej w tych wyborach. Jakie jest rozwiązanie? Porażka zawsze boli. Polacy tak dziś, w tym tygodniu, w niedzielę, jak i 5 lat temu dokonali wyboru zgodnego z zasadami demokracji. Wygrane wybory to zaangażowanie i ciężka praca każdego z kandydatów, praca sztabu, wolontariuszy, ale przede wszystkim decyzja wyborców. W 2015 r. to kandydat koalicji rządzącej wówczas, urzędujący prezydent Komorowski mimo zaplecza instytucji państwa, a dziś obecny kandydat Koalicji Rafał Trzaskowski przegrali wybory właśnie z Andrzejem Dudą. Dokonajcie więc państwo oceny, jakie znaczenie miały w całym procesie kampanii wyborczej instytucje państwowe. Kto decyduje o wygranej? Wyborcy. Czas pogodzić się z porażką.

Na pewno nie odpowiadały standardom państwa demokratycznego. Kilka faktów. Zaangażowanie telewizji publicznej. Przypomnę, w lutym br. Jacek Kurski o Andrzeju Dudzie mówił tak: Gdyby nie telewizja, nikt nie wiedziałby, kim jest ten człowiek. Oczywiście zaangażowanie 2 mld zł na przestrzeni tych miesięcy spowodowało, że dla telewidzów, dla widzów telewizji publicznej Andrzej Duda stał się pierwszym wyborem. Znacznie gorsza jest sytuacja związana z tym, co uczyniliście Rafałowi Trzaskowskiemu. Ta partyjna szczujnia zaangażowana na rzecz zohydzenia i obrzydzenia kandydatury Rafała Trzaskowskiego jest czymś, co musi być po prostu napiętnowane. Zaangażowaliście cały aparat państwa na rzecz jednego kandydata. Tu akurat zrobiliście wszystko, aby tam, gdzie można było zawieść, zawieść. Awaria systemu, żeby wyborcy nie dopisali się do spisu wyborców, w pierwszym dniu przed drugą turą wyborów czy kompromitujący przykład obwodu do głosowania w Splicie. Nie dało się utworzyć kilku obwodów do głosowania, kilku komisji? Trzeba było wszystkich zgromadzić w jednym miejscu? Przykładowe łapówki w postaci wozu strażackiego skierowaliście tylko do gmin do 20 tys. mieszkańców. A co, Polacy mieszkający w innych gminach są gorsi? Dlaczego tam nie było żadnego instrumentu zachęcającego do większej frekwencji? Odpowiedź jest prosta, jak się popatrzy na wyniki głosowania. A kto odbierał? Często radni. Jeden z radnych Krakowa trzyma (Dzwonek) czek na 19 mln zł, którego nikt nie widział i który nie ma żadnych podstaw prawnych. To czysta manipulacja. Dziękuję serdecznie. To, co trzeba powiedzieć o wyborach, które przeżyliśmy - to były wybory zgodne z literą prawa. I nie jest tak, jak mówił przedmówca, że te wybory były nieuczciwe. Nieuczciwe było to, że zachowania ze strony Koalicji Obywatelskiej, naszych przeciwników, nie tylko urągały godności człowieka, ale przede wszystkim poniżały każdą osobę, która reklamowała naszego obecnego prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudę. Nie mogę się również zgodzić z tym, że podważa się pracę urzędów, pracę ofiarną wszystkich pracowników.

Mówić można wszystko, ale jeżeli w legalnych, zaplanowanych zgodnie z prawem wyborach wygrywa kandydat, wtedy się składa z honorem gratulacje i przeprasza się za to, co się źle odbyło. Następna sprawa. Dlaczego te wybory się nie odbyły?

Dla mnie to jest skandal, że opozycja czyniła wszelkie zabiegi, żeby demokracja w Polsce nie wygrała. Mówię państwu, demokracja wygrała, wybory były przeprowadzone w sposób legalny, zgodnie z literą prawa, a jeżeli były jakieś wątpliwości, proszę, od tego są instytucje, gdzie można to zgłaszać. Wielki szacunek dla wszystkich pracowników, wolontariuszy, którzy.

Pan poseł Paweł Rychlik, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Wysoka Izbo! Jesteśmy po bardzo pracowitej kampanii prezydenckiej. Wszyscy kandydaci jeździli po Polsce, przekonując obywateli do swoich racji. Również prezydent Warszawy pan Rafał Trzaskowski jeździł do dziewięciu województw, w których to w wyniku awarii i przestoju działalności spalarni osadów przechowywane są osady pościekowe. Warszawa nie radziła sobie z utylizacją własnych osadów. czego konsekwencją było m.in. rozwożenie tych osadów po polach w innych województwach.

Osady te trafiały m.in. do Bogumiłowic w gminie Sulmierzyce, powiat pajęczański, województwo łódzkie. W większości tych miejsc Inspekcja Ochrony Środowiska zgłosiła szereg uwag i nieprawidłowości, m.in. w osadzie stwierdzono obecność salmonelli oraz innych bakterii, jaj pasożytów jelitowych. Można powiedzieć, że kurz powyborczy opadł, ale, panie pośle Nitras, syf został. Chciałem skierować pytanie do pana ministra. Bardzo serdecznie dziękuję. Nie za bardzo zrozumiałem tę sugestię w sprawie syfu, ale może. Nie chcę być złośliwy.

Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Zwolennicy Trzaskowskiego niszczą Polaków - to taki przykładowy, przykry, kuriozalny pasek, który pojawił się na ekranie w czasie głównego wydania Wiadomości w ostatnich godzinach kampanii, kolejnego wydania, które oczywiście w całości było poświęcone promocji jednego z kandydatów, czyli urzędującego prezydenta Andrzeja Dudy, i zohydzaniu drugiego z kandydatów, czyli kandydata opozycji Rafała Trzaskowskiego. Naprawdę nie potraficie inaczej? I mają dość m.in. tej obrzydliwej papki propagandowej, która każdego dnia wylewa się z telewizji publicznej. Co zrobili przedstawiciele rządu? Co zrobił minister kultury i dziedzictwa narodowego, który sprawuje w pewien sposób nadzór nad mediami publicznymi, by zapewnić kandydatom równy dostęp do mediów publicznych, który mamy zapisany w ustawie o organizacji kampanii wyborczej?

10 mln Polaków powiedziało, że ma dość waszej papki propagandowej, w tym ponad 60% najmłodszego pokolenia, które nie ogląda telewizji publicznej. Dziękujemy serdecznie za ten głos. Zapraszam uprzejmie pana posła Lecha Kołakowskiego z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. W związku z tym zapraszam uprzejmie pana posła Artura Łąckiego z Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska. Zdalnie? Ale nie przyfrunął. Proszę bardzo. Wysoka Izbo! Ja na temat tych kartoników, jak państwo z Platformy to nazywacie. Nie wiem, czy macie świadomość, że wasi samorządowcy też brali w tym udział. Byłem na kilku takich spotkaniach. W powiecie siedleckim tak się złożyło, że akurat zabrakło kartoników, dziwnym trafem, przypadek, nomen omen, dla prezydenta Siedlec pana Sitnika z Platformy Obywatelskiej. I odpowiedź pana prezydenta Sitnika: pana słowo mi więcej starczy niż kartonik. Dziękuję serdecznie. Pani poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Zapraszam panią poseł. Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Ten znakomity prezes telewizji publicznej was, drodzy państwo, coraz więcej kosztuje. Przed wyborami europejskimi i parlamentarnymi trzeba było dać z pieniędzy podatników 1200 mln. Studio wyborcze i jego szef, czyli pan prezes, kosztują. Ale teraz przed wyborami na prezydenta kandydatura Andrzeja Dudy kosztowała podatnika już 2 mld zł. Miliard dwieście było za mało. Razem, jak to policzyć, kochani, to 4 mld zł publicznych pieniędzy, poza funduszem sztabów wyborczych, poszło na kampanię Prawa i Sprawiedliwości. Wiecie, te 4 mld zł mogłabym przeliczyć na bardzo znaczący wzrost nakładów na onkologię. Gdybyście tych pieniędzy nie dawali telewizji publicznej, tobyście dzisiaj dali bon turystyczny każdemu emerytowi. A ponieważ poszło do studia wyborczego pod tytułem: telewizja rządowa, emeryci bonu nie dostaną. Dziękuję serdecznie, pani poseł. Chciałem państwu serdecznie podziękować za dzisiejszą współpracę. Jest moja koleżanka, pani wicemarszałek. A państwu dziękuję. Pan Dariusz Olszewski, Prawo i Sprawiedliwość. Pan poseł Cezary Grabarczyk, Koalicja Obywatelska. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie! To nie były uczciwe wybory. Przede wszystkim dlatego - o czym tu już była mowa - że została zatarta granica między państwem, między Rzecząpospolitą a partią. Tego w demokratycznym państwie prawnym czynić nie wolno. Konstytucja w sposób jednoznaczny w art. 7 stanowi, iż organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Kieruję pytanie: Jakie były podstawy prawne tego publicznego spektaklu wręczania łapówek, korupcji wobec samorządów i mieszkańców poszczególnych gmin? Jakie były podstawy prawne? Oczekuję, że odpowiedź padnie dzisiaj. Bo albo mieliśmy do czynienia z korupcją, albo mamy do czynienia z oszustwem. To w zależności od tego, czy te tekturki, tzw. czeki, będą miały pokrycie, czy też tego pokrycia nie mają. Albo korupcja, albo oszustwo. Czy ten rekonesans szefa rządu i ministrów z czekami po Polsce dał rezultat? Dał rezultat. Tam gdzie były odwiedziny z tekturkami, wzrosła frekwencja, w niektórych przypadkach aż o 19%, w wielu przypadkach o 10%. Czy ta sytuacja miała wpływ na wynik wyborów? Tak, w sposób oczywisty. Ale tego w demokratycznym państwie prawnym rządowi robić nie wolno. W każdym [[Dzwonek]] przypadku była bezpośrednia transmisja telewizyjna. A telewizja nie transmitowała ani jednego wiecu wyborczego Rafała Trzaskowskiego. Dziękuję bardzo, panie pośle. Pani poseł Teresa Pamuła, Prawo i Sprawiedliwość. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo! Wybory się skończyły, a państwo nie potraficie przegrać.

Jest tam inna ordynacja wyborcza, ale ja nie słyszałam do tej pory. Akurat miałam tę przyjemność i w tym czasie byłam w Stanach Zjednoczonych. Kiedy się położyłam spać, wygrywała Hillary Clinton. Wstałam rano - głosami elektorskimi wygrał Trump. Wiem, że podważano te wyniki, mówiono, że to Rosjanie mieli wpływ na to, że Trump wygrał. Ale Trump rządzi i ma wielu zwolenników. Tam mieliśmy 90-procentowe głosy na Dudę, na naszego prezydenta. I proszę zapytać: Czy te osoby, które głosowały na pana prezydenta Andrzeja Dudę, były manipulowane? Nie były manipulowane, panie pośle, na pewno nie. Tam żyją szlachetni, dobrzy ludzie, którzy głosują na wspaniałych ludzi, na wspaniałych. Na nic się zdadzą państwa krzyki.

Ja nie jestem zmanipulowana. A teraz się dowiaduję, że był zakaz. Nie wiem dlaczego. Pani Katarzyna. Bardzo proszę o spokój. Panie i Panowie Posłowie! Nie ma większego wstydu w sporcie, niż wygrać wtedy, kiedy się jest na dopingu. A to, co było z prezydentem Dudą, [[Oklaski]] to jest tak, jakby on startował na dopingu. To, z czym mieliśmy do czynienia, to był zorganizowany przemysł manipulacji. Zaczynał się na każdym szczeblu. Bardzo jasne: są dwie grupy wyborców, w których było wiadomo, że większość ma Duda. Jedna to są obywatele 60+, druga to są małe miasta. Dla jednych był sygnał RCB, który nie mówił o tym, żeby założyli maseczki i byli bezpieczni, tylko żeby poszli do wyborów, bo będą pierwsi w kolejce, a dla drugich były wozy strażackie w momencie, w którym nawet może nie być tam OSP, tak jak w jednej z miejscowości. Kolejna rzecz - telewizja publiczna. Telewizja publiczna, jeden wielki przemysł pogardy, który stosowaliście w stosunku do Rafała Trzaskowskiego. Przypomnijmy paski: Trzaskowski przeciwko katolikom. Czyje interesy reprezentuje Trzaskowski? Trzaskowski odbierze Polakom 200 mld. Ale są też paski o Dudzie. Ale są też paski o Dudzie: Duda obiecuje program propolski. Tłumy na spotkaniach z prezydentem Dudą.

Kolejna kwestia.

Poza wszelkim prawem, łamiąc prawo, wysłał do ludzi z KRUS-u. listy i ulotki Dudy. To jest przykład, który mieliśmy, manipulacji.

wiem i już jestem pewna, że temat tej informacji bieżącej z kłamliwą tezą jest próbą przykrycia nieprawidłowości, jakie miały miejsce w Warszawie, kiedy prezydent miasta, wiceprzewodniczący Platformy, chcący zresztą uchodzić za bezpartyjnego, zamiast zajmować się problemami Warszawy, prowadził swoją kampanię. Pokazujecie dobitnie, że nie szanujecie demokracji. Nie możecie pogodzić się z demokratycznym rozstrzygnięciem Polaków. Bojkotowaliście wybory 10 maja, blokowaliście realizację obywatelskiego przywileju i obowiązku. Straszyliście śmiercionośnymi kopertami, by po kilku dniach ochoczo zbierać podpisy na podmienionego kandydata. Przepraszam. Dziś po raz kolejny, po kolejnej przegranej znów kłamiecie i straszycie. A tymczasem według informacji Wód Polskich w czerwcu w czasie kampanii w Warszawie zrzucono ścieki komunalne do Wisły. Tutaj cytat: Zanieczyszczeń było tak dużo, że leciały terenem zielonym należącym do obszaru Natura 2000. To informacja prezesa Wód Polskich. Polacy, w tym mieszkańcy terenów nadwiślańskich, pytają, kto sprawował nadzór nad tym, co działo się w Warszawie, kiedy prezydent miasta zajmował się swoją kampanią wyborczą. Jeśli tak, to jakie? Polacy o to pytają? Zacznijcie wreszcie państwo i z Platformy, i z Koalicji Obywatelskiej szanować strażaków ochotników. Bo ja nie mogę się nie odnieść do tego, do tych słów, które tutaj padły, nie mogę jako druhna wspierająca OSP. Blisko 600 wozów ratowniczo-gaśniczych w tym roku zostanie przekazanych dla jednostek OSP w całej Polsce, także na Pomorzu. Zapytajcie tych druhów, którzy co roku dostają potrzebne im samochody, a których nie widzieli, nie mogli się doczekać za waszych rządów, kiedy, Platformo, rządziliście. Bardzo proszę, pani poseł Klaudia Jachira, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Chciałabym tylko pani posłance odpowiedzieć, zanim wyjdzie, że za czasów prezydenta Lecha Kaczyńskiego wszystkie ścieki trafiały do Wisły, ponieważ nie było wtedy jeszcze oczyszczalni. Ale teraz chciałabym wrócić do tematu naszej informacji bieżącej. Chciałam osobiście zobaczyć, jak wygląda głosowanie korespondencyjne za granicą, skąd biorą się liczne sygnały od naszych wyborców o nieprawidłowościach, dlatego zostałam mężem albo może raczej żoną w 93. komisji w ambasadzie w Berlinie. 24 godziny ta komisja obradowała, sprawdzała, liczyła te głosy. Naprawdę nie chcę pomyśleć, ile byśmy liczyli korespondencyjne wybory w Polsce. Ale przede wszystkim pragnę się dopytać o następujące nieprawidłowości. Dlaczego pod ambasadę w dzień wyborów przychodziły osoby, które dopisały się do spisu wyborców, ale w ogóle nie dostały przesyłki wyborczej, pakietu? Dochodziło do takich kuriozalnych sytuacji, że ludzie się sami organizowali i organizowali jakichś kurierów społecznych, żeby tylko jakoś te pakiety dostarczyć przed tą godziną 21. W komisji, w której obserwowałam wybory, 20 pakietów było zaadresowanych na nasze komisje, ale wyborcy znajdowali się w komisji obok, za ścianą i pani konsul odmawiała przeniesienia takich pakietów. Kto poniesie za to odpowiedzialność? Wreszcie, jak korespondencyjne wybory za granicą można uznać za równe, jeśli przez nierealne terminy, które państwo narzucili, wyborcy musieli płacić często po 15–20 euro na pakiet, by mieć nadzieję, że ten pakiet dojdzie na czas. Czy status materialny ma decydować o tym, kto może brać udział w wyborach? Tak naprawdę wymieniam pierwsze z brzegu nieprawidłowości, myśląc o nich i ich skali, tylko do mnie wpłynęło (Dzwonek) kilkaset takich skarg o wyborach za granicą. Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że zrobili państwo naprawdę wszystko, by utrudnić głosowanie Polonii w korespondencyjnych wyborach. Dlaczego? Pani poseł Agnieszka Górska, Prawo i Sprawiedliwość. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! A może, szanowni państwo, zapytamy, ile pieniędzy miasto stołeczne Warszawa, dzielnice miasta przelały na kontrakty, na konta niektórych warszawskich mediów na propagandę.

Czy to nie korupcja? Mimo to, mimo wydanych milionów polskich obywateli, mieszkańców Warszawy przegraliście wybory. Z tych mediów na pewno o tym się już nie dowiemy. Mogą one mieć teraz bezpośrednią motywację do obrony Rafała Trzaskowskiego, do przemilczania niewygodnych dla niego tematów: finansowania wybranych mediów i siania propagandy przy ich pomocy. To bardzo ważne, ponieważ to lokalne media powinny rozliczać władze samorządu. Z przerażeniem obserwuję, że w Warszawie jest niewielka ilość mediów, które nie boją się rozliczać z marnej działalności i trwonienia publicznych pieniędzy podczas kampanii wyborczej i nie tylko Rafała Trzaskowskiego i jego ekipy. To hańba. Dziękuję bardzo, pani poseł. Pan poseł Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pamiętacie państwo słynną grę na TikToku. Ministerstwo Cyfryzacji na promocję tej gry podczas kwarantanny wydało kilkaset tysięcy złotych. Kto był twarzą tej gry w czasie kampanii wyborczej? Andrzej Duda. Szanowni Państwo! Druga sprawa. Pamiętacie państwo uroczyste podpisanie w Żyrardowie na spotkaniu z seniorami ustawy dotyczącej tzw. trzynastej emerytury. Akademia w formule konwencji wyborczej? Kto zapłacił blisko 150 tys. zł za to wydarzenie? Zapłaciło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Chciałbym zadać pytanie, jak to się stało, że w czerwcu, 23 czerwca Państwowa Komisja Wyborcza wysyła - tutaj mam kserokopię - pismo do prezydenta miasta Tarnowa, w którym pan przewodniczący Marciniak pisze do prezydenta: Nieuzasadnione byłoby i niedopuszczalne przebywanie mężów zaufania oraz obserwatorów społecznych i międzynarodowych w lokalach komisji obwodowych utworzonych w zakładach leczniczych i domach pomocy społecznej, w których komisje powołane zostały na umotywowany wniosek osoby kierującej tą jednostką, wyłącznie spośród pracowników danej jednostki. Sprawdzamy te wyniki na stronie Państwowej Komisji Wyborczej. Pojawia się kilkaset przypadków w skali kraju, gdzie w zakładach opiekuńczo-leczniczych, gdzie przebywają osoby z niepełnosprawnością intelektualną, często bez jakiegokolwiek kontaktu, z bardzo zaawansowaną demencją czy chorobą otępienną, jest 100% frekwencji [[Dzwonek]] i 100% głosów na Andrzeja Dudę. Czy minister Szumowski występował do PKW w sprawie zakazu wejścia obserwatorów międzynarodowych, społecznych czy też mężów zaufania do tego rodzaju placówek stałego pobytu? Nie ma pana posła. Pan poseł Michał Gramatyka, Koalicja Obywatelska. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie! Jednym z najbardziej skrajnych przykładów wykorzystania zasobów państwa w służbie jednego tylko kandydata jest to, co państwo zrobili z jedną z najstarszych polskich spółek, z Pocztą Polską. Przypomnijmy, 23 kwietnia Poczta Polska wysyła do samorządów takiego maila, w którym żąda, prosi, żąda właściwie przekazania danych osobowych Polek i Polaków po to, żeby zorganizować tę farsę, którą planowaliście państwo na 10 maja. Niektóre samorządy przekazują te dane, ale nie wiadomo które i nie wiadomo ile rekordów, dlatego że ta informacja jest póki co ściśle strzeżoną tajemnicą. Od końca kwietnia usiłujemy się tego dowiedzieć, ale nikt nie chce nam odpowiedzieć. Podczas kontroli w siedzibie Poczty Polskiej udaje się nam ustalić, że ten mail jest wysłany na osobiste polecenie pana premiera Morawieckiego, że wiele samorządów odpowiedziało na tego maila i przesłało te dane, co więcej, że wiele samorządów przesłało te dane w formie plików otwartych, normalnym mailem, bez szyfrowania, bez hasłowania. Każdemu specjaliście od ochrony danych wrażliwych resztki włosów stają na głowie dęba, jak coś takiego słyszy. No i teraz moje pytania. Jak państwo wykorzystali te dane? Kto je widział? Kto je przetwarzał? Czy istnieje korelacja pomiędzy przekazaniem wam tych danych a tymi skandalicznymi i oszczerczymi ulotkami, które trafiły do skrzynek Polek i Polaków w czasie kampanii wyborczej i które mieszając z błotem jednego z kandydatów, wychwalały pod niebiosa drugiego? Tam nawet wizerunek najlepszej chyba osoby, jaką znam, pani marszałek Kidawy-Błońskiej, był pokazany w świetle negatywnym. ze wstydu podczas rozmowy z panem Thomasem Boserupem, czyli szefem misji OBWE w Polsce, który pytał mnie, czy w moim kraju zasoby państwa są wykorzystywane, żeby wspierać jednego kandydata. Można się pogodzić z porażką wyborczą, ale z porażką wyborczą, którą się ponosi w równej konfrontacji, a państwo oszukiwaliście na każdym etapie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani poseł Anna Kwiecień, Prawo i Sprawiedliwość. Wysoka Izbo! Platforma podobnie jak w 2015 r. nie może pogodzić się z faktem, iż w ciągu 5 lat pan prezydent zdobył zaufanie Polek i Polaków i w związku z tym Polacy ponownie wybrali pana prezydenta na to zaszczytne stanowisko. Wy państwo tak dużo mówicie o prawdzie, o tym, że ktoś kłamie. Szanowni państwo, no przecież ta kampania była wypełniona kłamstwami z państwa strony. Do 10 maja twierdziliście, że koperty będą zabijać, że macie kandydata, którego absolutnie nie podmienicie, a już 11 maja. To państwo potraktowaliście niezwykle instrumentalnie kobiety, wy, którzy zawsze tyle mówicie o kobietach. Najpierw potraktowaliście bardzo instrumentalnie panią marszałek, a potem. to już najbardziej haniebna sprawa.

Wykorzystanie życia tych kobiet to jest hańba z waszej strony.

Tej hańby nigdy z siebie nie zmyjecie. Nie wiem, czy zwróciła pani uwagę, że tych wyborów nie miała przeprowadzać Państwowa Komisja Wyborcza, a to nie jest zgodne z polską konstytucją i takie wybory nie powinny się odbyć. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Dzisiejsza informacja bieżąca poświęcona jest wysokiemu zaangażowaniu instytucji państwowych w proces wyborczy podczas ostatnich wyborów na prezydenta RP. Wszyscy z dużym zdziwieniem przyglądaliśmy się temu olbrzymiemu zaangażowaniu pana premiera Mateusza Morawieckiego oraz przedstawicieli Rady Ministrów. Oni tak się wyeksploatowali w tej kampanii wyborczej, że uznali, iż dzisiaj czas na odpoczynek i nie mają odwagi i chęci przyjść tutaj i stanąć przed Wysoką Izbą, aby odpowiadać na pytania. Szanowni Państwo! Informacja bieżąca to jest bardzo ważny punkt każdego posiedzenia Sejmu. Chcę zapytać: Gdzie są przedstawiciele rządu, którzy mogliby się odnieść do tych bardzo poważnych zarzutów? Rozumiem, że odpoczywają po ciężkiej kampanii wyborczej. Sama wasza telewizja publiczna informowała o tym, że premier Mateusz Morawiecki odbył aż 200 spotkań w 100 powiatach. Pytanie: Czy tak powinna wyglądać praca rządu podczas pandemii koronawirusa? Ale przechodząc do pytań, panie ministrze, będę pytała z uporem maniaka o wykorzystanie systemu alertu RCB w trakcie ciszy wyborczej. Obywatele byli oburzeni tym, że ten system został wykorzystany. Założenie tego systemu jest zupełnie inne. On ma informować obywateli o realnych zagrożeniach na danym terenie.

Będę dalej pytała, bo pana odpowiedzi mnie nie przekonały. Proszę odpowiedzieć na pytanie: Jaka była przesłanka do podjęcia decyzji o wysłaniu takiego komunikatu? Jakie wtedy występowało zagrożenie? Kto wydał decyzję o wykorzystaniu systemu alertu RCB? Czy pan premier był włączony w proces decyzyjny i czy istnieją procedury, które pozwalałyby w przyszłości uniknąć nadużywania tego systemu do celów politycznych?

Wysoka Izbo! Zaangażowaliście cały aparat państwa, żeby tylko przepchnąć na drugą kadencję swojego kandydata. Rząd nie pracował prawie miesiąc. Szef rządu w ciągu ostatnich tygodni zajmował się tylko kampanią na rzecz reelekcji Andrzeja Dudy i kłamał jak z nut.

Jacek Kurski w TVP dwoił się i troił, rozkręcając najobrzydliwszą kampanię w historii wolnej Polski. Zamiast pluralizmu, bezstronności i wyważenia mieliśmy w tych mediach zohydzanie i szczucie na Rafała Trzaskowskiego przez cały czas kampanii, a nawet podczas ciszy wyborczej. Nawet OBWE nie zostawiła na waszej brutalnej kampanii suchej nitki, zwracając uwagę na ksenofobię, homofobię i antysemityzm chociażby w mediach publicznych. Jeszcze PKW nie ogłosiła wyników, a już pojawiła się masa nieprawidłowości. Wyborcom z zagranicy staraliście się utrudnić oddanie głosu, jak tylko mogliście, bo wiedzieliście, że Rafał Trzaskowski miażdżył Dudę prawie w każdym kraju. W tej kampanii stawialiście na podsycanie niechęci do przeciwników politycznych i zachęcanie do agresji wobec różnych grup społecznych. Za pogłębiające się podziały w społeczeństwie po tych wyborach wy jesteście odpowiedzialni i wyłącznie wy za to będziecie odpowiadać. Jak wam nie wstyd? Pan poseł Dariusz Joński, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Wiele było wystąpień dotyczących telewizji tzw. publicznej, która poświęciła ogrom swojego czasu, atakując wszystkich kandydatów, z wyjątkiem pana Andrzeja Dudy. Nie było ani jednego materiału, chcę to bardzo wyraźnie podkreślić, ani jednego materiału, który byłby choć neutralny dla Rafała Trzaskowskiego bądź innych kandydatów, którzy ubiegali się o tę funkcję. To tylko pokazuje, z czym mamy do czynienia, jeśli chodzi o telewizję tzw. publiczną. Ale chciałbym się skupić na pewnym cytacie: Wybory sfałszowano. To początek drogi na Wschód. Drogie panie. W 2014 r. W ten sposób zmienia się ustrój w Polsce, bo państwo, gdzie fałszuje się wybory, nie jest już państwem demokratycznym. Wtedy nie sfałszowano. Ale te słowa wzięliście państwo sobie do serca jako cel do realizacji. Najgorsze jest, że prowadzicie nas na Wschód. Ale na szczęście 10 mln Polek i Polaków powiedziało wam: dość, i wcale tam nie chce iść.

Dziękuję bardzo. Ostatnie pytanie, pani poseł Marzena Okła-Drewnowicz, Koalicja Obywatelska. O telewizji tzw. publicznej, czyli propagandowej, na tej sali było już dużo, ale może konkretne przykłady.

Tego człowieka ułaskawił. Niech pani się douczy, co oznacza syndrom sztokholmski.

A on nie pomagał im, tylko m.in. telewizji propagandowej. Ta walka była po prostu nierówna.

Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu przedstawiciela wnioskodawców pana posła Borysa Budkę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Zero skruchy, zero pokory. Nie potraficie powiedzieć: przepraszam. Powinniście przede wszystkim przeprosić własnych wyborców, że w taki haniebny sposób ich traktujecie. Bo to, co robicie, to jest wielka pogarda dla intelektu zwykłych ludzi. My mamy wielki podziw dla każdego, kto wziął udział w tych wyborach. Mamy wielki szacunek dla każdego, kto oddał głos, bez względu na to, na kogo głosował. Ale absolutnie nie możemy się zgodzić na to, co wy wyczyniacie w Polsce. Zawłaszczyliście państwo, bowiem boicie się równej rywalizacji. Że wasz kandydat Andrzej Duda miał wtedy równy dostęp. Wy to wszystko zawłaszczyliście, bo to, czym się kierujecie, to jest olbrzymi strach, strach przed prawdą, strach przed tym, że król jest nagi. Boicie się powiedzieć o faktycznym stanie finansów publicznych. Obiecaliście czternastą emeryturę - nie ma tych pieniędzy.

Ale jesteście wyjątkowymi tchórzami. Dlaczego? Dlatego że boicie się prawdy, boicie się stanąć i powiedzieć, jaka powinna być Polska. Nie powiedzieliście niczego nowego w tej kampanii wyborczej, powtarzając ciągle kłamstwa i nieprawdę. Pan minister opowiada o wielkiej frekwencji, ale tysiące osób nie mogły wziąć udziału w święcie demokracji. Dlaczego? Bo jesteście nieudolni, bo po prostu nie chcieliście, żeby one głosowały.

My mówimy wyraźnie: Nie ma zgody na to, by rywalizować w ten sposób, by zawłaszczać państwo, by traktować instytucje publiczne jak własność jednej partii. Zrobiliście to z telewizją, próbujecie to zrobić ze służbami mundurowymi, zrobiliście to ze spółkami Skarbu Państwa. Wy mówicie o przeznaczaniu pieniędzy dla niektórych spółek, ale przecież to w poniedziałek Kurski zaatakował waszego premiera. Przecież to wy wydajecie pieniądze w tych firmach i nagle się oburzacie.

Tak traktujecie państwo. Jak dojną krowę, która zapłaci za waszą propagandę i fałsz. Te wybory nie były równe, te wybory nie były powszechne, ale przede wszystkim te wybory nie były uczciwe. bo wbrew temu, co wy mówicie, jesteście partią, która z uczciwością nie ma nic wspólnego. Zbudowaliście cały swój polityczny kapitał na kłamstwie. Zbudowaliście polityczny kapitał na kłamstwie o państwie w ruinie, na kłamstwie, jeśli chodzi o katastrofę smoleńską. Oszukiwaliście ludzi przez tyle lat, mówiąc o zamachach, mówiąc o państwie w ruinie.

I dzisiaj mieliście szansę stanąć tutaj i przeprosić Polaków, powiedzieć tak: Wygraliśmy nieuczciwie, sorry, wiecie, normalnie byśmy nie wygrali. Ale wy tego nie umiecie powiedzieć. Jesteście jak taki sportowiec na dopingu. Ta walka wyborcza wyglądała w ten sposób, że był ring otoczony ludźmi w amoku i w każdej przerwie Jarosław Kurski dodawał ten doping Andrzejowi Dudzie. Jest mi wstyd, że prezydent Rzeczypospolitej został tak wybrany, bo to będzie piętno na najbliższe 5 lat, bo brak tej demokratycznej legitymacji będzie skutkował tym, że głowa państwa będzie bardzo słaba.

Bardzo proszę o zabranie głosu sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji pana ministra Pawła Szefernakera. Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Rozumiem, że w pewien sposób wyjaśniłem tę kwestię merytorycznie. Jeżeli chodzi o te pytania, które padły, o zdrowie i życie Polaków - tak, proszę państwa, jesteśmy w czasie epidemii. Chciałbym przypomnieć, że te SMS-y były w taki sam sposób wysyłane jak te, które były wysyłane w kwietniu, w marcu tego roku.

Pan, panie pośle Nitras - ta pana śmieszna maniera mówienia: młody człowieku, o młodym człowieku. Niech pan to zostawi, bardzo proszę, dla swoich koleżanek, kolegów z Młodych Demokratów, a w polskim parlamencie może się pan do mnie zwracać: panie ministrze lub panie pośle. Odnosząc się do tego, co pan powiedział na mój temat z tej mównicy, mogę jedynie powiedzieć, że właściwie właśnie pan, szczególnie pan po tej kampanii Rafała Trzaskowskiego i pana roli w tej kampanii nie jest w stanie mnie obrazić, naprawdę. Jedyne, co jest pan w stanie, to mnie rozśmieszyć. W trybie sprostowania pan poseł Sławomir Nitras. Szanowny Panie Ministrze Szefernaker! Pan swoją wypowiedzią dokładnie udowodnił, że to jakiś kaprys pana Brudzińskiego spowodował, że pan jest ministrem, a nie pana kompetencje. Przecież my tu od godziny mamy zarzuty dotyczące telewizji, roli administracji państwowej, 200 spotkań wyborczych premiera Morawieckiego za pieniądze publiczne, tego, że schrzaniliście specjalnie wybory za granicą, bo tam Trzaskowski wygrywał, i w tych państwach, w których są wyborcy Trzaskowskiego. Zrobiliście w Bułgarii lokal wyborczy w Sofii. W Złotych Piaskach, w Słonecznym Brzegu są setki tysięcy Polaków, a wy w Sofii zrobiliście, 600 km od wybrzeża, bo wam nie zależało na tych głosach, bo wiecie, że ci Polacy głosują na kogoś innego. Pan jest człowiekiem niedojrzałym. A wie pan, dlaczego pan jest ministrem? Chodzi o to, żeby tu stawał człowiek poważny, który, gdy są zarzuty dotyczące wykorzystywania mediów publicznych np. w kampanii, do tego się odniesie, [[Dzwonek]] a pan tego nie potrafi. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych pana ministra Piotra Wawrzyka. Panie i Panowie Posłowie! Pojawiło się tu kilka omówień opinii OBWE na temat wyborów, więc ja państwu przeczytam dosłowny fragment: Wszystkie szczeble administracji wyborczej kontynuowały wywiązywanie się ze swoich obowiązków w sposób profesjonalny pomimo trudności związanych z głosowaniem podczas pandemii COVID-19. Zarówno kandydaci, jak i władze zachęcali wyborców do aktywnego głosowania w drugiej turze. W ograniczonej liczbie lokali wyborczych odwiedzanych przez obserwatorów proces głosowania oraz liczenia głosów odbywał się w sposób sprawny i dobrze zorganizowany, a obostrzenia sanitarne były ściśle przestrzegane. W związku z tym wybory zostały przez OBWE uznane za w pełni demokratyczne.

Dlaczego wracały?

Awaria systemu wyborczego. Zwracam uwagę, że nie jest tak, że system wyborczy prowadzi Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Infrastruktura techniczna, która zapewnia jego funkcjonowanie, i sam system są prowadzone przez operatora zewnętrznego, jednego z dużych operatorów telekomunikacyjnych, i to po jego stronie leżała wina w odniesieniu do awarii, która miała miejsce. ale zwracam uwagę, że to jest kurort, w którym przyszło na wybory w drugiej turze cztery razy więcej wyborców niż w pierwszej, niemniej oczywiście każdy wyborca, który się tam pojawił, otrzymał możliwość oddania głosu.

Jeżeli chodzi o Berlin, pani poseł, zwracam uwagę, że zgodnie z decyzją władz niemieckich wybory mogły się odbyć wyłącznie w drodze korespondencyjnej, w związku z tym niemożliwe było też dopisanie się do spisu.

Co do Bułgarii, panie pośle, tak samo. Przepraszam, ale proszę się zwrócić do władz Bułgarii, dlaczego zgodziły się na otwarcie lokalu wyborczego tylko w Sofii. To nie była nasza decyzja. A gdyby pan wiedział, gdyby pan miał doświadczenie w tym zakresie, którego panu brakuje, toby pan wiedział, że odbywa się to w drodze not, które wysyła się do władz, informując o chęci przeprowadzenia wyborów. i w tej samej drodze poszczególne kraje odpowiadają na nasze noty. Tak się odbywa to w dyplomacji.

Tutaj padło bardzo dużo zarzutów pod adresem m.in. telewizji publicznej i generalnie systemu medialnego w Polsce.

także inne telewizje mają taki sam obowiązek, bo on jest wpisany bardzo wyraźnie w koncesji. Koncesja mówi bardzo wyraźnie każdej telewizji, że każda telewizja powinna równoważyć wszystkie strony w zakresie informacji. Proszę państwa, pierwszy raz od wielu lat, przez ostatnie kilka lat wreszcie mamy sytuację, kiedy infosfera jest zrównoważona. Mamy pluralizm. jedną, jedynie słuszną narrację innych stacji telewizyjnych. I telewizja publiczna skutecznie to robi. Dziękuję państwu.

Informacja o wpływie interpelacji i zapytań oraz odpowiedzi na nie dostępna jest w Systemie Informacyjnym Sejmu. Protokół posiedzenia będzie wyłożony do przejrzenia w Sekretariacie Posiedzeń Sejmu.